Szczęść Boże! Wysoka Izbo! Proszę skończyć z tą farsą. To jest farsa - powoływanie się na niedoskonałości jednej z sieci telefonicznych w sytuacji, w której te obrady są zamknięte, tak jak cały kraj zamknięty jest w kwarantannie, na własne życzenie aktualnego układu władzy. Skończcie z reglamentacją dostępu do tej sali, otwórzcie nam komisje sejmowe, zespoły parlamentarne. Nie uniemożliwiajcie wprowadzenia czynnika społecznego, naszych rodaków, do prac Sejmu.

Proszę z tym skończyć. Nie udzielam panu głosu, panie pośle. Bardzo pana proszę, żeby pan przychylił się do tego, co ustaliło Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, czyli reprezentanci nas wszystkich, żebyśmy przystąpili do pierwszego czytania ważnego rządowego projektu, na który wszyscy czekają. Nie możemy głosować, ponieważ nie wszyscy posłowie mają dostęp. Ja? Tak, panie pośle, pan. Pan, panie pośle, tak, oczywiście, że tak.

Mam inną propozycję, dobrze? Bardzo państwa proszę.

Za chwileczkę jeszcze raz poproszę o sprawdzenie, ilu posłów się zalogowało. Jeżeli się okaże, że w dalszym ciągu mamy spore braki, to za zgodą Konwentu Seniorów przystąpimy do rozpatrzenia punktu 2., czyli sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Kluby zadeklarowały, że ich przedstawiciele są przygotowani do tego punktu. W międzyczasie będę ciągle sprawdzała, czy nam posłów przybyło, czy nie ma tego problemu, i wtedy wrócimy do porządku dziennego. Tak, czyli następna byłaby informacja rządu, ta, o którą wnioskowała Koalicja Obywatelska. Zwracam się do wszystkich państwa posłów obecnych tu, na sali, w innych salach, a także zdalnie łączących się z nami o to, żeby wcisnęli jeszcze raz dowolny przycisk, żebyśmy sprawdzili, jaką mamy w tej chwili liczbę posłów, którzy biorą udział w głosowaniu. Bardzo proszę.

Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad punktami porządku dziennego. Proszę państwa, w takim razie państwo chyba nie zrozumieliście, co mówiliśmy, co ustalaliśmy wspólnie, że wnioski formalne będą głosowane wtedy, kiedy zniknie problem, tak? Dobrze, możemy i tak zrobić. W takim razie. Dokończę tylko, pan pozwoli, tę formułkę. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie występowania suszy na terenie Polski, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia Sejmu będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Chciałam tylko zwrócić uwagę, proszę państwa, że ten komunikat może ulec zmianie w związku z przesunięciem związanym z tą sytuacją, czyli proszę śledzić komunikaty, o której godzinie odbędzie się posiedzenie komisji, bo to może ulec zmianie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Zwracam się z wnioskiem formalnym o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem uzupełnienia porządku obrad o informację premiera w sprawie przygotowań do wyborów prezydenckich. Czego się boicie? Tego, że OBWE mówi, że wybory będą niedemokratyczne, czy decyzji, którą ogłosił przewodniczący PKW, mówiąc, że nie będą to wybory wolne? Namawiacie samorządowców do łamania prawa, karty wyborcze drukujecie tak, jak w „Piłkarskim pokerze”, a sprawy dotyczące legalności wyborów prokurator umarza w ekspresowym tempie. Ze święta demokracji robimy farsę. W imię Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wzywam, abyśmy dzisiaj albo na najbliższym posiedzeniu, czyli w ciągu tych 3 dni, przegłosowali ten wniosek, a wszyscy, którzy nie będą chcieli współpracować - nie chcą przeprowadzić uczciwych wyborów. Proszę bardzo, drugi wniosek, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Wysoka Izbo!

W mediach elektronicznych czytać można wypowiedź pana marszałka Terleckiego, który występuje albo jako - ośmielam się wykluczać taką perspektywę - współsprawca problemów z połączeniami, albo też jako prorok mniejszy, który wyprorokował, że kogoś może tam zabraknąć, ktoś się może nie połączy. Przeczytajcie państwo, co pan marszałek Terlecki. Może pani marszałek zachęci Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby sprawdziła, czy istotnie zachodzi okoliczność, ta pochlebna dla pana marszałka, że pan marszałek zaledwie przewidział, a nie doprowadził do takich problemów z połączeniami. Wniosek o odroczenie. Pan poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska - PSL - Kukiz15.

Właśnie przed chwileczką się dowiedziałam, że jest taka sytuacja.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Również w trybie art. 184 regulaminu Sejmu wnoszę w imieniu klubu Koalicja Polska o zarządzenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów celem, o czym uprzedzałem na poniedziałkowym zdalnym posiedzeniu Konwentu, rozszerzenia porządku obrad o rozpatrzenie uchwały zgłoszonej już prawie miesiąc temu przez nasz klub, wzywającej rząd Rzeczypospolitej Polskiej przez Sejm do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Krótkie uzasadnienie. W dokumencie, w projekcie ustawy, który będziemy dzisiaj rozpatrywać, czyli tzw. tarczy 3, w uzasadnieniu dotyczącym zmiany trybu powoływania składu Krajowej Rady Prokuratorów rząd pisze: aby wybory mogły się odbyć w jak najbezpieczniejszy sposób, czas na ich przeprowadzenie ustalono na 90 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ostatni wniosek, pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Proszę o uzupełnienie porządku dziennego o projekt poselski, który zgłosiła Koalicja Obywatelska. Ten projekt dotyczy testowania pracowników domów pomocy społecznej, innych placówek opieki stałej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek prywatnych oraz hospicjów. Ten projekt, szanowni państwo, jest już złożony. Pani marszałek ma ostatnio taką tendencję, żeby wprowadzać do porządku obrad nawet projekty, które nie mają numeru druku sejmowego. Apeluję do pani marszałek o uzupełnienie porządku obrad o projekt Koalicji Obywatelskiej, który jest złożony. On dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w placówkach opieki stałej, dotyczy również bezpośrednio pensjonariuszy tych placówek. Uważamy, że co tydzień wszyscy pracownicy w tych najbardziej narażonych miejscach, jakimi są miejsca pobytu stałego osób w wieku senioralnym, powinni być testowani. Jeżeli otwieramy, pani marszałek, 4 maja galerie handlowe, żłobki czy też instytucje kultury, to apeluję, żeby następne posiedzenie Sejmu odbyło się w normalnych warunkach, nie Sejmu zdalnego, który jest, jak widać, bardzo kruchy, ale w normalnych warunkach fizycznej obecności posłów w gmachu Sejmu. Dziękuję bardzo.

W sali 118 jest już obsługa, która problem rozwiązuje. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druki nr 269 i 321) Proszę pana posła Marka Suskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Przepraszam, ale dobiegłem z drugiej sali, gdzie głosowałem. W tej maseczce trochę trudno złapać oddech. Można zdjąć. Będę mógł złapać oddech. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji do rządowego projektu zmiany ustawy - Prawo energetyczne, druki nr 269 i 321. To jest projekt dotyczy ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej wobec takiej infrastruktury. Jest to, szanowni państwo, projekt dostosowujący polskie prawo do prawa Unii Europejskiej. Jest to też związane z tym, że Polska wnioskowała, aby tego typu rozwiązania zostały przyjęte w Unii Europejskiej. Będzie to obejmować wszystkie połączenia gazowe z krajami Unii Europejskiej, czy są to kraje Unii, czy spoza Unii, czy jest to rurociąg, gazociąg rosyjski łączący z Unią Europejską, czy są to polskie gazociągi łączące z Litwą, Słowacją czy innymi państwami z nami sąsiadującymi. Jest to poprawka dotycząca promocji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi o wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z tym, czy wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy przyłączeniowej jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucji stanowi podjęcie decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy, co uniemożliwiałoby spełnienie tzw. efektu zachęty.

Konsekwencją poprawki będzie zmiana nazwy proponowanej ustawy. Szanowni Państwo!

Zgłoszono szereg różnego rodzaju uwag, ale generalnie zdecydowana większość była za tym, żeby ten projekt wraz z poprawkami poprzeć.

W mojej opinii, cytuję, zaproponowana zmiana jest zasadna i będzie służyła rozwojowi kogeneracji opartej o paliwa gazowe w kraju. Projekt nowelizacji został wcześniej uzgodniony z Urzędem Regulacji Energetyki. To rozwiewa wątpliwości, jakie były zgłaszane na posiedzeniu komisji. W związku z tym bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tego projektu, gdyż jest on potrzebny polskiej gospodarce. Dziękuję, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał ten projekt wraz z poprawką. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Rozmawiamy dzisiaj o implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2019 r. Sprawozdawcą był pan premier, europoseł Jerzy Buzek.

Efekt tej dyrektywy dla Polski, szczególnie z punktu widzenia gazociągu Nord Stream 2, jest pozytywny. Po pierwsze, zaniechali wdrożenia tej dyrektywy tak szybko, jak się da, przekroczony został termin, dlatego że dyrektywa mówi, że państwa członkowskie powinny to implementować do 24 lutego.

Te regulacje były mocno kwestionowane na forum europejskim oraz - co za tym idzie i co bardzo ciekawe - ten dwugłos pomiędzy przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w rządzie i w Parlamencie Europejskim.

Możliwe, że bałagan jest wewnątrz rządu, pomiędzy Ministerstwem Energii a pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Przy okazji tej implementacji prawa europejskiego pojawia się zmiana ustawy o promowaniu energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji. Bardzo dziwna sytuacja, bo w żaden sposób nie odnosi się ona do dyrektywy. Czy to oznacza, że polski rząd ma jakieś nowe propozycje odnośnie do rozwiązania problemów wynikających z błędnych decyzji ministra Tchórzewskiego co do budowy bloku energetycznego w Ostrołęce i teraz próbuje ten blok ustanowić na gazie? Może warto byłoby na ten temat trochę dłużej w polskim parlamencie porozmawiać, jak rząd to widzi. A tutaj po cichutku, tylnymi drzwiami nowelizuje się ustawę, która nijak się ma do wspomnianej dyrektywy. Ta dyrektywa, jej wprowadzenie pokazuje też, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo często lubi mówić, politycy Prawa i Sprawiedliwości lubią mówić o tym, że tak naprawdę instytucje europejskie chodzą na pasku Niemców. Warto więc podkreślić, że dokładnie ta dyrektywa interesy niemieckie, szczególnie te związane z Nord Stream 2, mocno nadwyręża. Zadaje to też kłam tezie, jaką przez wiele lat politycy Prawa i Sprawiedliwości prezentują, że Komisja Europejska, instytucje europejskie tylko i wyłącznie działają pod dyktat państwa niemieckiego. Nasuwa się pytanie, jak polski rząd ma zamiar oddziaływać na Komisję Europejską w sytuacji, kiedy do regulatora niemieckiego wpłynie wniosek Gazpromu o wyłączenie inwestycji Nord Stream 2 z działania tejże dyrektywy, bo przypominam, że te inwestycje, które zostały zakończone, choćby w części europejskiej, przed majem 2019 r., mają prawo uciec od tej dyrektywy, która bardzo jasno opisuje, jakie są obowiązki właściciela tego gazociągu, i pozwala na dostęp stron trzecich. Krótko mówiąc, nie wie lewica, co robi prawica.

Dziękuję bardzo.

Zamykam więc - to nie jest głosowanie - sprawdzanie, ilu nas jest. Poproszę o zabranie głosu pana posła Dariusza Wieczorka, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jest to wprost implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która została przyjęta w 2019 r. Tak jak pan przewodniczący Suski mówił, rzeczywiście jest to dyrektywa, która jest bardzo korzystna i porządkuje cały ten system w skali Unii Europejskiej. Natomiast rodzi się pytanie, czemu tak późno implementujemy dyrektywę do polskiego prawa. Argumenty były takie: a to były wybory, a to ukonstytuował się polski rząd, a to trafiła się pandemia - w związku z czym nie mieliśmy czasu, żeby to realizować. Zwracam uwagę na to, że Prawo energetyczne - i w ogóle energetyka - jest ważną dziedziną, w związku z czym potrzebne są bardzo szybkie działania ze strony polskiego rządu po to, żebyśmy czegoś nie przegapili, jeżeli chodzi zarówno o gaz, jak i o prąd. Rodzi się więc pytanie, czy rzeczywiście polski rząd ma pod kontrolą całą branżę energetyczną. Przypomnę, że w planach polskiego rządu, w planie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na I kwartał tego roku znajdowała się kwestia dotycząca zmiany Prawa energetycznego, nie tylko w tym obszarze, o którym dyskutowaliśmy i który jest tutaj podany, ale zdecydowanie i znacznie szerzej.

Oprócz Prawa energetycznego potrzebne są również w tym zakresie zmiany wielu innych ustaw, chodzi chociażby o kwestię dotyczącą rynku mocy i ustawy o rynku mocy. Mamy nowelizację ustawy o elektromobilności i uruchomienie w ogóle tego procesu. Na razie zmieniamy tylko terminy wejścia, nie rozwiązując rzeczywistych problemów. Bardzo ważna sprawa to kwestia prowadzenia w ogóle inwestycji sieciowych gazowych i energetycznych, a więc kwestia dotycząca ustawy o korytarzach przesyłowych, dyskutowana już w poprzedniej kadencji, przez wiele lat.

Wiem, że w planach pracy komisji i planach rządowych ten zapis się znajduje, natomiast przypomnę, że pracujemy nad tą polityką od 2018 r., a jest rok 2020.

To świadczy o tym, że mamy problemy, jeżeli chodzi o moce wytwórcze, mamy problemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie energetyki. W związku z tym dzisiaj panuje w energetyce duży chaos organizacyjny i chaos inwestycyjny. Co jest tego powodem? Po pierwsze, przyjmowanie ludzi powiązanych tylko i wyłącznie z ugrupowaniem rządzącym, którzy nie mają pojęcia o gazownictwie i nie mają pojęcia o energetyce, biorą pensje i - mówiąc krótko - często są jak słynny yeti: wszyscy wiedzą, że są zatrudnieni, ale nikt ich w tych przedsiębiorstwach nie widzi. Po drugie, brak kompetencji w zarządzaniu.

To są decyzje, które powodują, że mamy bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o inwestycje, takie jak chociażby elektrownia Ostrołęka, kwestia przejęcia Orlenu przez Energę. To są rzeczy, o których warto dyskutować. Reasumując, chcę powiedzieć, że klub Lewica poprze proponowany projekt ustawy, natomiast apelujemy do rządu o to, ażeby - mówiąc krótko - zabrał się za pracę w sektorze energetycznym. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak, zdalnie. Bardzo proszę.

Musimy chwilę poczekać, bo się

Mamy jakieś problemy techniczne, jeśli chodzi o połączenie z panem posłem. W związku z tym przechodzimy do pytań. Zamykam listę chętnych do zadawania pytań. Jako pierwsza zada pytanie pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja. Przepraszam bardzo.

Panie pośle, do sekretariatu przyszła informacja, że pan w ogóle zrezygnował z wystąpienia, ale skoro pan przyszedł, bardzo proszę. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pan poseł Robert Winnicki. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy powstał dlatego, że nie działa w Unii Europejskiej podstawowa zasada, która powinna konstytuować tę wspólnotę, tę domniemaną wspólnotę. Chodzi o solidarność, solidarność państw w obliczu najważniejszych, największych wyzwań. Nie ma tej solidarności, ponieważ największe państwo, hegemon Unii Europejskiej, Republika Federalna Niemiec wbrew interesom wszystkich państw Europy Środkowej forsuje kolejne gazociągi, Nord Stream 2, przedkładając swój interes narodowy ponad interesy państw mniejszych. To jest fakt. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy epidemia koronawirusa uświadamia nam, jak wiele zależy od państw narodowych i kiedy to państwa narodowe właśnie w Unii Europejskiej walczą o swoje interesy, o swoje bezpieczeństwo, walczą z epidemią, to jest fakt, który uświadamia nam, że podstawowe założenie, na którym oparta jest Unia Europejska, po prostu nie działa. Od kilku lat, od ładnych kilku lat trwa walka o to, żeby wymusić na Niemcach solidarność w kluczowej kwestii, kwestii bezpieczeństwa energetycznego, a oni prą zgodnie ze swoim interesem narodowym, który postrzegają sprzecznie z interesem państw Europy Środkowo-Wschodniej. To po pierwsze.

To po pierwsze. Po drugie, to również zadaje kłam całej retoryce Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która chwali się od wielu lat, jak to dobre ma relacje właśnie na Zachodzie, właśnie w Brukseli, właśnie w Berlinie. Otóż okazuje się, że te dobre relacje z Brukselą czy z Berlinem są tylko w jedną stronę, tzn. dzisiaj Polska jako podwykonawca gospodarki niemieckiej, dzisiaj Polska jako żyrant przez lata, od traktatu lizbońskiego co najmniej, polityki centralistycznej Republiki Federalnej Niemiec - to jest wszystko w jedną stronę. To jest wszystko w jedną stronę, ponieważ kiedy chodzi o nasze interesy, to musimy na Niemcach wymuszać. Musimy na Niemcach wymuszać i oczywiście zobaczymy jeszcze, z jaką skutecznością. Trzecia kwestia to kwestia energetyki i kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Szanowni państwo, zwracam tutaj uwagę, że wszelkie działania zmierzające do dywersyfikacji gazowej są potrzebne, pożądane i generalnie co do zasady popieramy w tym zakresie działania rządu. Dywersyfikacja energetyczna.

Dzisiaj Polska potrzebuje realnej dywersyfikacji i myślenia nie tylko o tym, jak się uniezależnić od Moskwy, jak się uniezależnić i zabrać ten pistolet szantażu, ten szantażystowski pistolet gazowy ze strony Moskwy, ale również ze strony Zachodu, jak się uniezależnić również od tej drugiej strony, ponieważ nie wiemy, jakie wyzwania polityczne, gospodarcze czy militarne zgotuje nam przyszłość. Dzisiaj to jest wyzwanie polskiej polityki zagranicznej i do tego również wzywamy rząd, żeby tę politykę wielowektorową, tak na gruncie dyplomacji, jak i na gruncie polityki surowcowej, realnie prowadził. Dziękuję. Dziękuję bardzo.

Przepraszam za te kłopoty, ale przez kilka minut pracowaliśmy dość intensywnie ze służbami, aby uzyskać to połączenie.

Otóż zabierając głos. Panie pośle, przepraszam.

Teraz chyba dobrze, bo ten pogłos się skończył. Teraz w ogóle pana posła nie słychać. Jeszcze raz witam i przepraszam wszystkich, ale tak to jest z techniką. Słychać mnie? Proszę mówić. Teraz bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.

Panie pośle, proszę śmiało mówić. Coś się nam tutaj psuje. Chcę powiedzieć tak: dyrektywa.

Wypowiadaliśmy się publicznie na ten temat, znamy stosunek Unii Europejskiej. Już połowa krajów implementowała tę dyrektywę, w tym również strona niemiecka. Niemcy implementowali to do swojego prawodawstwa, z tym że 2 dni po przyjęciu przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa projektu tej ustawy, po debacie w komisji, mogliśmy spotkać się z komentarzem ze strony Rosji, która wręcz naciska, nalega na stronę niemiecką, aby Niemcy wyłączyły się z obowiązku tej dyrektywy. To jest bardzo niezrozumiałe i bardzo niepewne. W tym przypadku wydaje mi się, że jest to bardziej intencyjna dyrektywa, ale każdy z nas życzyłby sobie, żeby jednak doszło do pełnego przestrzegania tej dyrektywy. Naciski i interesy Rosji znane są w Europie. Stosunki. Coś mi przerwało.

Ważne jest, że dzisiaj Europa zaczyna dywersyfikować dostawy gazu, jeżeli chodzi o różne kierunki. Myślę, że w przyszłości to, co zostało już kilka lat, a może i kilkanaście lat temu zapoczątkowane, przyniesie skutki.

Będziemy popierać ten projekt.

Myślę, że to też jest korzystne. Wysoki Sejmie!

Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy wystąpienia klubowe. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Porozmawiajmy o energii. Na wczorajszym spotkaniu Rady Unii Europejskiej ds. energii minister Kurtyka mówił o potrzebie bezpieczeństwa dostaw energii czy większego udziału energii odnawialnej w Polsce. Ale tyle teoria w ustach ministra klimatu. Niestety w praktyce, zamiast negocjować miliardy euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, minister klimatu szukał drogi do uzależnienia naszej energetyki od zagranicznego, drogiego gazu. Minister mówił: dla Polski gaz stanowi najszybszą dostępną ścieżkę umożliwiającą ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza. Panie ministrze, czy inwestycje gazowe naprawdę są najszybszą i najtańszą ścieżką ograniczenia emisji i budowania niezależności energetycznej? Absolutnie nie są. Nie mamy polskiego gazu. Importowany gaz jest dużo droższy niż polski wiatr i polskie słońce.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo!

Jednakże polski rząd nie zadbał o to, aby w odpowiednim czasie wdrożyć, zaimplementować przepisy, które dają możliwość polskim firmom energetycznym skorzystania z ulg, ale także stworzenia wspólnego rynku wewnętrznego handlu gazem. Moje pytanie jest następujące: Czy z racji tego, że zostały przekroczone terminy wdrożenia implementacji, polscy przedsiębiorcy, polskie firmy energetyczne nie utracą ulg, zwolnień z niektórych obowiązków? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Jeśli już nie utracą, to dlaczego zgodnie z zapisami ustawy polskie firmy mają zaledwie 7 dni (Dzwonek) na złożenie wniosku o ubieganie się o zwolnienie?

Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! To już zostało wspomniane: w lutym minął czas transpozycji przepisów tej dyrektywy do porządku krajowego. Jak zwykle Prawo i Sprawiedliwość pokazało szacunek dla prawa europejskiego i spóźniło się z implementacją. Nawet w takiej kwestii nie potrafiliście na czas implementować przepisów. Ten dyskutowany projekt ustawy, który, jak słusznie zauważył sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek, będzie popierany przez Lewicę, to jest tylko wycinek czegoś znacznie większego, czyli po prostu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Ta polityka musi powstać przy współudziale wszystkich sił parlamentarnych w Polsce. To jest niezwykle ważne, by później mogła być realizowana niezależnie od tego, czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy rządzi Lewica.

Czy będzie to realizowane ponad politycznymi podziałami? Kiedy będą konsultacje społeczne i kiedy odbędzie się szeroka debata publiczna na temat tego dokumentu, który ciągle jest w powijakach i ciągle jest tylko projektem? I pani poseł Beata Maciejewska, klub Lewica. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

To są ogromne spadki cen. Dotyczy to także innych spółek i koncernów energetycznych: PGE, firm Tauron i Enea. Czy to nie jest powód, żeby zastanowić się, dlaczego polska energetyka tak mocno traci i czy rzeczywiście nie powinniśmy dzisiaj wdrożyć całościowej koncepcji energetycznej, całościowego planu, o którym zresztą już wcześniej mówiliśmy? Pracujemy na odcinkach. Pracujemy tak, jakbyśmy kładli tory na odcinku 500 m mniej więcej co 3 km i pomiędzy jednym a drugim odcinkiem nie ma żadnego połączenia. Chciałabym wiedzieć, czy i w jakim terminie wreszcie zorganizujemy (Dzwonek) naszą politykę energetyczną w taki sposób, żeby miała ona ręce i nogi. Przypomnę, że nie mamy dzisiaj nawet ministerstwa energii. Kolejne pytanie zada pani poseł Katarzyna Ueberhan, Lewica. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed nami wspólne cele, ale tez wspólne wyzwania, takie jak ograniczenie emisyjności, jak zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, ale również konkurencyjności cen czy zagwarantowania faktycznego wyboru każdemu odbiorcy energii bez względu na to, czy jest to przedsiębiorca, czy jest to obywatel.

Pan poseł Janusz Cichoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.

Szanowna pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówimy o przepisie europejskim, przepisie, który będzie miał, jak możemy przeczytać w ocenie skutków regulacji, korzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku gazu ziemnego, zwiększy konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, także polskiej gospodarki, zwiększy wreszcie bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski. To wymierne korzyści, ale w tym OSR-ze zakładacie państwo, że nie będziecie prowadzili ewaluacji tego projektu, że nie będzie OSR-u ex post. Że boicie się, że czarno na białym będzie widać, jakie rzeczywiście korzyści płyną z przynależności Polski do Unii Europejskiej w takim drobnym tylko fragmencie.

Zapraszam. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Na te pytania nie mamy odpowiedzi, ale pojawia się dzisiaj jasny punkt w wykonaniu naszego premiera i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Otóż własną inicjatywą doprowadził do przygotowania regulacji europejskiej, która eliminuje monopol Gazpromu na ceny przesyłu.

Ta dyrektywa jest przejawem solidarności, za co należą się ogromne podziękowania panu premierowi Buzkowi. Do tego stopnia, że nawet Niemcy zgodziły się pod presją na wdrożenie tej dyrektywy.

Pan poseł Grzegorz Braun, koło Konfederacja. Wysoka Izbo! Frazes przywracania suwerenności w dziedzinie energetycznej króluje na tej sali.

Superminister, a może nawet superpremier Obajtek byłby mile widziany, bo jeżeli chodzi o wszystko, co się w tej branży dzieje, to są sprawy, na które nie tylko w urzędzie Rady Ministrów, w Pałacu Prezydenckim, ale może nawet i przy Nowogrodzkiej niektórzy są za krótcy, a pan prezes Obajtek wie, co robi. Pytanie, czy wiedział, co robi, kiedy doprowadzał do przejęcia Energi przez Orlen, co stawia polski sektor energetyczno-paliwowy wobec ryzyka wrogiego przejęcia. Proszę państwa, warto na tej sali więcej na te tematy mówić. Już pika automat, pani marszałek zabiera mi głos, więc kończę, kłaniając się.

Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Implementacja dyrektywy europejskiej w sprawie Prawa energetycznego jest bardzo ważna, bo zapewnia pewność prawa dla uczestników rynku. W przypadku wprowadzania tych zmian konieczne jest jednak zadanie pytania o dywersyfikację źródeł energii, która powinna polegać na zdecydowanym zwiększeniu udziału w polskim miksie energetycznym energii ze źródeł odnawialnych kosztem zmniejszenia udziału węgla kamiennego i brunatnego.

W perspektywie będzie to jeszcze większy udział. Proszę zatem o odpowiedź na piśmie na pytanie, jakie rząd planuje zmiany legislacyjne pozwalające na rozbudowę źródeł zielonej energii, kiedy one będą przedłożone Sejmowi, a także czy planowane są wysłuchania publiczne w tej sprawie. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj oczekiwałbym, że rząd również przedstawi polską energetykę, jeśli chodzi o przyszłość co do węgla, zwłaszcza zielonej energii, bowiem trzeba wykorzystać fundusze europejskie. Nie trzeba się od tego odcinać, trzeba walczyć o fundusze europejskie, bo tu się nic nie zmieni. Ceny prądu w Polsce są bardzo, bardzo wysokie. Niepokojący jest fakt, że my tej energii bardzo dużo importujemy. Proszę państwa, dzisiaj w globalnej gospodarce nie wystarczy machać szabelką. Dzisiaj trzeba rozmawiać zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze politycznej, a to pokazuje dobre kontakty w Unii Europejskiej i to (Dzwonek), że nawet trudne projekty są do przeprowadzenia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kolejne pytanie zada pan poseł, minister Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Oczywiście cieszymy się z tego, że pan przewodniczący Jerzy Buzek w sposób lojalny poparł nasze postulaty na forum Unii Europejskiej, i oczywiście do tej lojalności zachęcam, żebyście się państwo jako politycy Platformy Obywatelskiej uczyli od pana prof. Jerzego Buzka. A co do relacji polsko-niemieckich to rzeczywiście jest tak, że 10 września 2019 r. Polska wygrała przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej spór z Komisją Europejską dotyczący monopolizacji gazociągu OPAL, czyli lądowej odnogi gazociągu Nord Stream, i chcę powiedzieć, że Niemcy rzeczywiście zaskarżyły do wyższej instancji ten wyrok, podważając zasadę (Dzwonek) solidarności energetycznej. Jeżeli chcecie pomóc Polsce, poproście waszych kolegów z CDU, żeby nie podważali zasady solidarności energetycznej i nie sądzili się z Polską. Pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie przedstawicielom rządu. Z czego wynika tak wysoka cena energii z polskiego węgla?

W jakiej formie Unia Europejska złamała konwencję z Kioto, która pokazywała, że Polska więcej pochłania dwutlenku węgla dzięki lasom, rolnictwu i zielonym terenom, niż emituje?

Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! A mianowicie do Gdańska zawinął kilka dni temu największy masowiec w historii polskich portów, przywiózł węgiel z Kolumbii. Sprowadzamy ze wszystkich kontynentów węgiel, poza Antarktydą. Chciałbym pana ministra zapytać dokładnie o ten transport i o ten węgiel, który został sprowadzony z Kolumbii. Chciałbym również przypomnieć Wysokiej Izbie, że w ciągu ostatnich 2 lat sprowadziliśmy do Polski ponad 35 mln t węgla kamiennego o łącznej wartości 14 mld zł. Najwięcej, bo blisko 23 mln t - Rosja. Czy to jest właściwy kierunek polityki energetycznej?

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Informuję, iż lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W imieniu rządu głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan minister Ireneusz Zyska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić stanowisko rządu w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Parę faktów, nawiązując również do pytań, które szanowni państwo, panie posłanki i panowie posłowie, byli uprzejmi zadać. To przede wszystkim informacja o tym, że jest to inicjatywa rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pani premier Beaty Szydło i później pana premiera Mateusza Morawieckiego. To rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości zabiegał na forum Unii Europejskiej o wdrożenie i przyjęcie tej dyrektywy.

Nawiązując do wypowiedzi mojego szanownego kolegi, pana ministra Janusza Kowalskiego, trzeba powiedzieć, że bardzo doceniamy rolę pana prof. Jerzego Buzka, który jako przewodniczący komisji do spraw energii w Parlamencie Europejskim popierał starania rządu polskiego i dzięki temu te prace zakończyły się sukcesem. 17 kwietnia 2019 r. dyrektywa została przyjęta. Natomiast odnośnie do zarzutów, które były tutaj formułowane, dotyczących wdrożenia dyrektywy nie w terminie, to chciałbym poprosić szanownych państwa parlamentarzystów. Tutaj słyszałem też wypowiedź pana posła Borysa, który z dużą dozą pewności stwierdzał, że Polska jako ostatni kraj. Otóż informuję Wysoką Izbę, że do tej pory, do dnia dzisiejszego sześć państw Unii Europejskiej implementowało dyrektywę gazową. Polska jest 7. krajem, który w tej chwili tej implementacji dokonuje, tak że nie jesteśmy ostatni, jest całkiem nieźle. Natomiast opóźnienie wynika z tego faktu, że ta ustawa jest w przedłożeniu rządowym i jako taka wymaga pełnej ścieżki legislacyjnej, a dodatkowo jako implementacja dyrektywy - uzgodnień. Musimy to uzgodnić, jak państwo wiedzą. Pan minister Paweł Poncyljusz ma doświadczenie w pracach rządu, więc powinien pamiętać, że wymaga to uzgodnień z Komisją Europejską w zakresie tekstu ustawy, treści ustawy. Było zbyt mało czasu do wyborów parlamentarnych na jesieni ub.r., aby dokonać pełnej implementacji, z kolei procedura jest tak skonstruowana, że po wyborach musimy tę procedurę rozpocząć od nowa.

Odpowiadając na kilka kluczowych pytań, które tutaj zostały sformułowane, to bardzo ciekawe jest stwierdzenie pana posła Roberta Winnickiego. Rzeczywiście trzeba zauważyć, że Unia Europejska ma problem z podstawową wartością, jaką jest solidarność w wymiarze europejskim.

Kilka słów na temat dyrektywy. Mianowicie przede wszystkim daje ona uprawnienia stronom trzecim do włączenia się do ewentualnego gazociągu transgranicznego, a także wyłącza możliwość takiego rozwiązania, że właściciel gazociągu jest jednocześnie dostawcą gazu, tak jak Gazprom w przypadku (Dzwonek) Nord Streamu. Ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Ten gazociąg, regulacja tego gazociągu będzie podlegała prawu europejskiemu. Chcę też podkreślić, że wszystkie gazociągi transgraniczne, które przez Polskę w tej chwili przebiegają, są regulowane prawem europejskim. Bardzo przepraszam, mamy mało czasu. Bardzo słuszna uwaga jest również pana posła Marka Suskiego, przewodniczącego komisji, dotycząca złamania przez Komisję Europejską czy szerzej przez Unię Europejską protokołu z Kioto.

Też inne obciążenia zostały nałożone na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ale co niesłychanie istotne, proszę państwa, co warto, żeby opinia publiczna wiedziała: Polska jako strona, jako państwo członkowskie mogła powalczyć o odstępstwa, o derogacje w zakresie tych warunków, które zostały narzucone przez Unię Europejską w ramach systemu ETS, ale polityka rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a konkretnie pana premiera Donalda Tuska i pani premier Ewy Kopacz, niestety była niezgodna z polskim interesem i doprowadziła do nadmiernych, niewspółmiernych obciążeń polskiej gospodarki w stosunku do warunków, jakie np. uzyskała Francja czy też Niemcy.

Nie chciałbym mówić w tej chwili o szczegółach, bo jest to projekt, ale strona polska zaproponuje nowe rozwiązanie w zakresie regulacji dotyczącej systemu ETS, tak aby on był bardziej sprawiedliwy i bardziej efektywny. Na tę chwilę tyle. Dziękuję bardzo, panie ministrze. O głos poprosił sprawozdawca komisji pan poseł Marek Suski. Zapraszam pana, panie pośle. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom, którzy pracowali nad tym projektem, ponieważ mimo różnic politycznych wszyscy byliśmy zgodni, że jest to rozwiązanie korzystne dla naszego kraju. Mam nadzieję, że zdecydowana większość go przyjmie. Rządowi też życzę jego szybkiej realizacji. Ale poprawek nie ma, więc na tym zakończę. Dziękuję państwu za współpracę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję wszystkim państwu biorącym udział w dyskusji. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. W tej chwili zarządzam 10-minutową przerwę, po której przystąpimy do zapowiedzianych wcześniej głosowań. Dziękuję bardzo.

Tak że przerwa - 10 minut, szanowni państwo. Dziękuję.

Wznawiam obrady. W związku z tym bardzo proszę wszystkich państwa posłów obecnych na sali plenarnej, poza salą plenarną i łączących się z nami zdalnie o naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w celu sprawdzenia kworum. Bardzo proszę.

Proszę o wyniki.

Stwierdzam kworum. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem do zastosowania art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu do projektu ustawy z druków nr 344 i 344-A sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Kto z pań i panów posłów jest za skróceniem terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Wniosek o przerwę zgłoszony w imieniu klubu Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 przez posła Jacka Protasiewicza nie zostanie poddany pod głosowanie, ponieważ jest tożsamy z wnioskiem o przerwę i został już przegłosowany, natomiast wniosek o uzupełnienie porządku dziennego zgłoszony przez posła Michała Szczerbę nie będzie poddany pod głosowanie, ponieważ jest to wniosek nieregulaminowy. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 344 i 344-A) Proszę ministra - członka Rady Ministrów pana Łukasza Schreibera o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

To jest tak naprawdę dalsze uzupełnienie naszej tarczy antykryzysowej. Cieszę się, że Wysoka Izba będzie mogła nad tym projektem obradować. Chciałbym przedstawić ten projekt w następujący sposób, żeby pokazać, że faktycznie mamy konkretne zmiany dotyczące ułatwień dla przedsiębiorców, czy może szerzej: ułatwień w ratowaniu miejsc pracy. Po 10 takich najważniejszych spraw z tego projektu ustawy pozwolę sobie krótko omówić, a poza tym kilka innych fragmentów, które wykraczają poza ten stan rzeczy. Chciałbym zwrócić uwagę, że projekt zakłada, iż dla samozatrudnionych, tak jak to po poprawkach w Senacie przyjęła Wysoka Izba, jest możliwość przechodzenia na postojowe bez maksymalnej kwoty przychodu na poziomie trzech średnich krajowych, czyli ok. 15 600. Teraz wprowadzamy taki impuls, żeby zachęcać do aktywności, żeby oni rzeczywiście dalej mogli kontynuować pracę.

Jeżeli ten dochód nie jest wyższy niż 7 tys. zł, a przychód został przekroczony nawet o 15 600, to będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u. Tutaj też ważna uwaga, która się z tym wiąże: to nikogo nie wyklucza, żadna grupa, która dotąd została objęta tym zwolnieniem, nie będzie wykluczona. Druga sprawa.

Trzecia zmiana to zwolnienia z ZUS-u dla tych, którzy korzystali z ulgi na start i zaczęli działalność gospodarczą. Za kwiecień i za maj zostaną oni objęci tym zwolnieniem. Czwarta zmiana, techniczna, ale dla niektórych dość istotna, to zniesienie przepisu blokującego księgowanie korekt dokumentów rozliczeniowych na kontach płatników.

Następna, ósma zmiana dotyczy organizacji (Dzwonek) pożytku publicznego. Te organizacje dotąd, jeżeli korzystały ze środków z PFRON-u na dofinansowanie dla pracowników, nie były objęte możliwością skorzystania z szeregu mechanizmów zawartych w tarczy antykryzysowej. Teraz chcemy to zapewnić.

Dziesiąta sprawa, o której można powiedzieć, to wydłużenie terminów z tytułu sprawozdań, obowiązków informacyjnych, np. zakres rejestru bazy danych odpadowych - to jest przedłużone do końca roku. To jest te 10 spraw dla przedsiębiorców. Zacznę pewnie od jednej z najważniejszych. To są kwestie dotyczące lichwy, a tak naprawdę antylichwiarskie zapisy.

Teraz wprowadzamy kolejne mechanizmy.

Owszem, będzie mogło nastąpić przeniesienie własności nieruchomości, ale kwota pożyczki, którą się bierze, będzie musiała wynosić minimum 80% wartości nieruchomości, która zostanie określona przez rzeczoznawcę.

Zabezpieczenie tej sytuacji to oczywista korzyść dla obywateli, zwłaszcza w tym trudnym czasie, wyeliminowanie szeregu patologii.

Druga sprawa to odmrożenie gospodarki.

Wprowadzamy jednocześnie mechanizm złotówka za złotówkę.

Eliminujemy także to.

Wprowadzamy przepisy, które będą zobowiązywać operatorów do informowania abonentów o tym, że ich aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, natomiast przed automatycznym przedłużeniem operatorzy będą informować o możliwych sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Tu zwłaszcza myślimy rzecz jasna o osobach starszych, żeby zapewnić im takie możliwości. Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Wprowadzamy także dodatkowe, nowe wymagania, jakie powinny być uwzględniane podczas opracowania założeń dotyczących postępowań selekcyjnych. Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania jest unieważnienie ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji. Nie mają wszystkie charakteru epizodycznego, ale są ważne.

Wsparcie sektora drzewnego.

Nic takiego. 100% uposażenia dla żołnierzy, dla funkcjonariuszy na takich samych zasadach jak dla medyków, w przypadku gdy są oni w kwarantannie. To jest doprecyzowanie tych zapisów, bo od początku taka była intencja, doprecyzowanie także tych zapisów, poprawienie, które znoszą te decyzje, przywracają tak naprawdę te decyzje sądowo-administracyjne i ich bieg. Trzecia kwestia to rozszerzenie w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami możliwości procedowania w ramach tzw. rozprawy odmiejscowionej, to w sądach. To także dopuszczenie możliwości rozpoznania apelacji w postępowaniu cywilnym wniesionych przed dniem 7 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w szerszym zakresie. To także uproszczona możliwość przenoszenia sędziego do innego wydziału na podstawie nieprawomocnego podziału czynności.

Wysoka Izbo! Kończąc, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proszę pamiętać, kiedy państwo będziecie być może mówić o tych sprawach czy przypominać inne, o dwóch sprawach: o tym, co było w ostatnich dniach, mówię o uchwale Rady Ministrów, która zakończyła na tym etapie legislacyjnym proces tarczy finansowej, a więc o tych 100 mld zł dla polskich przedsiębiorców na pożyczki, na subwencje umarzalne w 75% - to lada dzień wejdzie w życie, mamy już zgodę, notyfikację Komisji Europejskiej - a także o tym, co będzie, czyli drugim projekcie ustawy, który lada moment trafi do Wysokiej Izby, którego wnioskodawcą jest minister rozwoju, pani premier Jadwiga Emilewicz, który z kolei rozszerzy i da kolejne możliwości przedsiębiorcom, tam się znajdzie ta tzw. tarcza samorządowa. Kończąc, chciałem prosić Wysoką Izbę o pilne procedowanie tego projektu. Dziękuję pani marszałek za włączenie go do programu dzisiejszych obrad. Jak państwo widzicie, jest tu naprawdę szereg dobrych, korzystnych zmian dla obywateli. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Andrzej Kosztowniak. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pozytywnego oczywiście, dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z druków nr 344 i 344-A, wraz z rządową autopoprawką do tego druku. Projekt ustawy stanowi kontynuację i uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ma na celu wprowadzenie kilku czy kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne. Jak pan minister zauważył, dzieli się to de facto na dwie grupy, z jednej strony na grupę finansową, a z drugiej strony jest to wsparcie odnoszące się przede wszystkim do systemu procedowania w wielu obszarach. Bardzo istotne są ułatwienie i pomoc dla przedsiębiorców i umożliwienie dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu, której działalność pozwoli na ograniczenie problemów przedsiębiorców związanych z pozyskaniem finansowania. Szanowni państwo, pozyskanie finansowania dzisiaj jest jednym z większych problemów dla przedsiębiorstw. Bardzo istotną rzeczą jest rozszerzenie zwolnień, umożliwienie skorzystania ze zwolnień z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia, w sytuacji gdy ich przychody były wyższe niż 300% prognozowanych przychodów przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. Wydaje się, że jest to znakomity ukłon w stronę tych wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mających relatywnie wysokie przychody w swojej działalności, ale dochodowość tych interesów, biznesów jest relatywnie niższa. Myślę, że to jest spory ukłon w stronę przede wszystkim małego handlu na terenie naszego kraju, ale również dużej części świadczonych usług. Jest to wprowadzenie terminów czy też wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków sprawozdawczych, o których była mowa. Ponadto ustawa wprowadza dalsze regulacje sprowadzające się do ograniczenia skutków pandemii dla przewoźników kolejowych i autobusowych, była już o tym mowa. Jest to pomoc dla rolników i producentów rolnych, ochrona i pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, m.in. wspomniane już podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 900 zł z 800 zł, wraz z wprowadzeniem zasady złotówka za złotówkę. To także rozszerzenie katalogu spraw, których załatwienie będzie możliwe drogą elektroniczną, co jest bardzo istotne w odniesieniu do procedowania nie tylko przed urzędami, ale w dużej mierze również przed sądami, umożliwienie wniesienia pisma do sądu powszechnego poprzez użycie platformy ePUAP w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii, umożliwienie dokonania doręczenia przez sąd za pomocą platformy ePUAP, usprawnienie i wsparcie w zakresie szkolnictwa wyższego i edukacji, o których była mowa, i usprawnienie działania sądu w trakcie epidemii za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie te propozycje jak najbardziej wychodzą naprzeciw wszystkim apelom, prośbom, które płynęły z bardzo wielu środowisk gospodarczych i społecznych. Wydaje mi się, że z jednej strony będziemy luzować pewne procedury z racji tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ale z drugiej strony zostały przygotowane bardzo konkretne instrumenty. Myślę tutaj o instrumentach finansowych, przede wszystkim zwolnieniach, które wniosą dużo dobrego dla polskiego biznesu, nie tylko tego największego.

Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej pan poseł Jarosław Urbaniak.

Wysoka Izbo! Kolejny projekt ustawy niby-dotyczący epidemii, niby-dotyczący walki ze skutkami tej epidemii i kryzysu gospodarczego. Piękny tytuł, piękne uzasadnienie, jak do tej pory cudowne słowa ze strony PiS-u, a w środku prawie nic. Oczywiście jest kilka listków figowych, ale nam przedstawiono prawie 200 stron przepisów, a tak naprawdę to, co dobre w tej ustawie, zmieściłoby się na jednej stronie. Tak naprawdę to, co dobre w tej ustawie, to realizacja naszych postulatów - Koalicji Obywatelskiej, które zgłosiliśmy przy poprzednich projektach ustaw. A jeśli zobaczyć, co w tym jest, to nie ma poza tym nic. Po pierwsze, brakuje najważniejszych postulatów. Nie ma słowa na temat badań testowych dla służb medycznych. Dzisiaj, 29 kwietnia wiemy, że najlepiej walczy się z epidemią tam, gdzie są obowiązkowe i systematyczne badania dla służb medycznych. Nadal nie ma uwolnienia handlu w niedziele, nadal nie ma uwolnienia pieniędzy pochodzących z VAT, z podzielonej płatności. To są pieniądze polskich podatników. Pozwólcie chociaż polskim podatnikom płacić wynagrodzenia z tych pieniędzy. Oczywiście nie ma słowa na temat ruchu przygranicznego. To jest walka z kryzysem? Nie ma słowa o specjalnych strefach ekonomicznych. Jeśli nie poluzujecie przepisów, tysiące firm w specjalnych strefach ekonomicznych zbankrutuje. A co mamy? No nie wolno tak, nie ma trybu przyspieszonego, panie ministrze.

To jest także złamanie regulaminu Sejmu, no ale to u was jest normą od 2015 r. A co jest? Wszędzie tam są ukryte brudy. Tak jak w poprzednich ustawach, tak i tutaj robicie wrzutki, dzięki którym kryjecie brudy. Jedno słowo zamienione jak słynne „lub czasopisma” Jak zamienicie słowo „prawne” na „faktyczne”, rząd będzie miał lepszy, łatwiejszy dostęp do danych osobowych polskich obywateli. Co ona ma wspólnego z epidemią?

Ano tylko wydłuża kadencje nominatów Ziobry np. w Krajowej Radzie Prokuratorów. Ustawa o telekomunikacji. Pan minister tutaj mówił, że teraz będzie transparentny wybór, a właściwie nabór na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Otóż nie. W tej procedurze brakuje Senatu, który do tej pory tu był. No bo PiS nie ma większości w Senacie. I taki nowo wybrany prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostanie nowe prawa, bo jak się wczytamy, to się okaże, że w szczególnych przypadkach, nie wiadomo jakich, taki prezes może ograniczyć prawa odbiorców usług telekomunikacyjnych. I to będzie walka z kryzysem: wyłączanie Polakom telefonów komórkowych i Internetu. To jest walka z kryzysem? Nie, to jest walka z opozycją. Prawo o transporcie kolejowym.

Dlaczego luzujecie także sposób wydawania pieniędzy z Funduszu Kolejowego? Patrząc na to, że znieśliście kary za niestosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, ja się domyślam dlaczego. Prawo łowieckie. Ano to, że tu mówicie, że zarząd Polskiego Związku Łowieckiego może podejmować decyzje o wydatkowaniu pieniędzy. Tylko chcę wam powiedzieć, że zarząd już podjął decyzję wbrew kołom łowieckim i zabrał te pieniądze. Przepisy antylichwiarskie. Brzmi bardzo dobrze, a naprawdę to jest walka SKOK-ów z firmami pożyczkowymi. No i Karta Nauczyciela. Dlaczego ogranicza się Kartę Nauczyciela i daje szeroko otwartą furtkę ministrowi, żeby tę kartę ograniczyć? Co mają wspólnego awanse zawodowe z tym, żeby przeprowadzić egzaminy maturalne lub egzaminy ósmoklasistów? No to jest po prostu skandal. Znowu zwykłą ustawą wprowadzacie nowy podatek w trybie nadzwyczajnym.

Teraz w imieniu klubu Lewicy pan poseł Krzysztof Gawkowski. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mija drugi miesiąc od kryzysu, jego początku, a rząd cały czas nie przedstawił porządnego planu wyratowania polskiej gospodarki, polskich pracowników. Wstyd. Wstyd, panie premierze. Rząd zamiast planu ratowania gospodarki i rozmrażania gospodarki ma plan, ale jest to plan przeprowadzenia wyborów. Lewica przedstawiła porządny program antykryzysowy. Podaliśmy jak na tacy: świadczenie kryzysowe, czyli 2600 zł dla każdego, kto stracił pracę albo zamknął firmę, podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł, zwolnienie z rat kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych. Wy na to wszystko: nie trzeba, za dużo, mamy inne pomysły. Przyjrzyjmy się zatem tym pomysłom. Co chcecie? Premier mówi: możliwość zwalniania pracowników przez e-mail, obniżanie pensji pracownikom o połowę, wyrzucanie na bruk pracowników, którzy pracują na drugim etacie. To jest wasza prawdziwa tarcza. Powiedzmy sobie szczerze, to jest lunatykowanie we mgle. Gracie ze społeczeństwem w rosyjską ruletkę i na wszelki wypadek załadowaliście cały magazynek. Bieda coraz częściej zaczyna gościć w polskich domach i rodzinach, a wy zamykacie oczy. Z tygodnia na tydzień proponujecie coraz gorsze rozwiązania, coraz bardziej szkodliwe, niebezpieczne dla społeczeństwa. Chcecie przerzucić koszty kryzysu na obywateli, pracowników, przedsiębiorców. Robicie wszystko, aby lekarstwo, które fundujecie polskiej gospodarce, było gorsze od samej choroby. I co najgorsze, milionom ludzi, którzy tracą pracę, którzy zamykają firmy, którzy nie mają za co godnie żyć, pokazujecie gest pani Lichockiej. Tak, gest pani Lichockiej.

Teraz proszę o głos panią poseł Monikę Falej, również klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Przykro mi to mówić, ale projekt tej ustawy to nie tarcza 3.0, a nerwowa próba wmówienia, że robicie wiele dla poprawy losu Polek i Polaków, a tak naprawdę robicie wiele hałasu o nic. Szumnie mówicie o tarczy, a co ona przedstawia? A przy okazji znowu nic nie mówicie, nic nie proponujecie dla pracowników, jakby zupełnie nie istnieli. A nie, jednak pan nie zapomniał: dzięki tarczy 2.0 łatwiej będzie właśnie obniżyć im pensje, zwolnić ludzi z pracy, chociażby osoby w wieku emerytalnym. Myślałam, że to ma polegać na czymś innym. A cała reszta ustawy, tzw. tarczy? Połowa zapisów nie ma nic wspólnego z epidemią. To jest worek z łatami na wasze dziurawe ustawy, chaotyczna zbieranina, a nie realny projekt pomocowy. Bo jak na walkę z koronawirusem ma wpłynąć zapis dotyczący wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez udziału Senatu? Co ma do rzeczy wspieranie Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego i możliwość powoływania nowych jego oddziałów czy też absurdalny pomysł, żeby minister edukacji narodowej mógł sobie dowolnie zmieniać ustawę - Karta Nauczyciela rozporządzeniem? Niektóre zmiany może i mają sens, są rozsądne, jak te w Kodeksie karnym. Można by się nad nimi nawet zastanowić, ale one nie pomagają w walce z koronawirusem. Podejrzewam, że prace nad tą ustawą wyglądały po prostu tak: zadzwonił pan do swoich ministrów, kazał im coś wymyślić, a ci w popłochu zaczęli urządzać sobie koncert życzeń i przedstawili swoje propozycje od Sasa do Lasa. Jest chaotycznym zapisem istniejącego już prawa, a nie realnym pakietem pomocowym. To, co dzisiaj nam przedstawił rząd, to nie tarcza, a mozaika wątpliwych propozycji, nad którymi powinno się głosować z osobna, jak nad poprawkami zapisów poszczególnych ustaw. Nie na to czekały miliony Polek i Polaków. Czas się kończy, panie premierze. Czas na poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków. Przyznajcie, że nie dajecie rady, póki jeszcze nie jest za późno. Lewica w komisji będzie składać merytoryczne poprawki.

Jak pan dalej będzie nas tak zapowiadał, jak przed chwilą, to marszałek Zgorzelski wszystkich posłów PiS-u będzie zapowiadał jako posłów Porozumienia. To po pierwsze. Kolejny akt tragifarsy pt. dziurawa i spóźniona tarcza antykryzysowa, pisany w przerwach pomiędzy wprowadzaniem wyborów pocztowych na wzór bawarski. Mieliście czerpać i przywieźć do Polski reparacje niemieckie, a czerpiecie z głosowania korespondencyjnego w Bawarii, które rozniosło koronawirusa. W przerwach próbujecie stworzyć pomoc dla pracowników i przedsiębiorców, po raz kolejny nieudolną. Dlaczego w innych państwach przyjęto jedną tarczę antykryzysową, która działa, funkcjonuje, a tutaj trzecia odsłona, która nie spełnia nawet obietnic składanych 3 tygodnie temu przez premiera Morawieckiego. 3 tygodnie temu wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polskiego pan premier Morawiecki wyszedł i powiedział o funduszu płynności. Powiem szczerze, ucieszyliśmy się, ucieszyli się pracodawcy w Polsce, związki pracodawców. Tylko co się z tym stało? Była zapowiedź, piękna konferencja prasowa. W PR-ze, w TikTokach jesteście mistrzami, ale w realnym działaniu już nie. Czytaliśmy 2 dni temu w „Rzeczpospolitej”, mówił o tym pan poseł Gawkowski: zwolnienia przez e-mail, ograniczenie czasu pracy, przez to ograniczenie wynagrodzenia i zwolnienie pracownika przez e-mail. To jest ratowanie miejsc pracy? Tarcza antykryzysowa dla tych wybitnych specjalistów miała być od tego, żeby ratować miejsca pracy. Wam się wszystko pomieszało. Wy w tym pędzie na oślep, na ścianę, bez hamulców do wyborów korespondencyjnych nie jesteście w stanie odróżnić ochrony miejsc pracy od zwalniania pracowników przez e-mail.

Chcecie wprowadzić opłaty od korzystania z Netfliksa i innych platform, na których można oglądać filmy i seriale. W momencie, kiedy Polacy zostali zamknięci w domach, był to często jedyny sposób rozrywki, uatrakcyjnienia dnia. Tylko wiecie, kto za to zapłaci? Polacy, nasi rodacy, nie wielkie koncerny, bo przerzucą te koszty. Na to nie może być naszej zgody. Chcecie obciąć nadgodziny pracownikom, funkcjonariuszom Policji. I taka nagroda, że nadgodzin dla nich nie będzie? To jest wsparcie, to jest solidarność? Z nami nie chcieliście solidarności. Powiem szczerze, że jedną rzeczą po raz kolejny mnie zaskoczyliście. Myślałem, że po 5 latach jest to już prawie niemożliwe, ale wasze zdolności są jednak nieograniczone. Ja się z nim spieram, polemizuję, ja z nim konkuruję, ale wy mówicie, że go popieracie. On kilkanaście dni temu mówił: trzeba zwolnić wszystkich pracowników, pracodawców z ZUS-u, umorzyć składki ZUS-owskie. Super, dobrze, też byśmy się z chęcią pod tym podpisali. Co prawda, jak my to mówiliśmy, to uważaliście to za licytację, za koncert życzeń ze strony opozycji. Interes pracowników i pracodawców jest dla nas ważniejszy, więc z chęcią chcieliśmy zgłosić te poprawki w Senacie. Tam je zablokowaliście. Dla was to nic nie znaczy, co powie Andrzej Duda. On jest wam potrzebny tylko do jednego i te wybory utrwalające władzę są wam potrzebne tylko do jednego: żeby akceptował wasze decyzje. Co trzeba zrobić? Plan dla Polski i trzy podstawowe rzeczy. Fundusz płynności natychmiast, pieniądze dla firm, żeby zapłacili pracownikom, żeby kupili towary, żeby mogli realizować usługi. Druga sprawa: dobrowolny ZUS na stałe, nie tylko czasowo, bo to jest w momentach kryzysowych konieczne, w momentach, kiedy jest lepiej, by była możliwość skorzystania, żeby nie zadusić polskich firm. I rzecz bardzo ważna: premia dla bohatera.

Pan poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Otwieramy projekt ustawy, która jest trzecią wersją tarczy antykryzysowej, i w art. 15 znajdujemy przepisy, które nie mają nic wspólnego z walką z kryzysem. Mianowicie rząd w art. 15 wprowadza nowy podatek bez żadnej dyskusji, bez żadnych konsultacji, bez żadnego namysłu, bez żadnej logiki. W uzasadnieniu możemy się dowiedzieć, że będzie on odprowadzany do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, a więc nawet nie w celu walki z kryzysem, nie w celu ochrony zdrowia, właściwie nie wiadomo w jakim celu. Gdyby Państwowy Instytut Sztuki Filmowej nie miał pieniędzy, to przecież premier, skoro sytuacja budżetowa była tak doskonała, z pewnością by dosypał, ale nie trzeba było dosypywać. Teraz jest wprowadzany nowy podatek. Na pierwszym miejscu Ipla, na drugim Player, na trzecim Amazon, na czwartym CDA, na piątym Netflix, Apple. Czy kogoś nam na tej liście brakuje? Oczywiście brakuje dwóch największych platform internetowych, które zgarniają prawie wszystkie budżety reklamowe w Internecie. Oczywiście są to dwie firmy amerykańskie. Czy to, co robi rząd, to podatek cyfrowy, o którym tyle mówił? Czy w tej chwili bocznymi drzwiami wprowadza jakąś wykastrowaną wersję w sposób wylobbowany przez panią ambasador? Czy o to chodzi? Dlaczego rząd postanowił opodatkować akurat to, za co Polacy sami płacą, czyli filmy, które sobie opłacą? Dlaczego rząd nie zdecydował się opodatkować tego, co jest dostarczane bezpłatnie, i tych firm, które zgarniają większość budżetów reklamowych? Jestem przeciwnikiem wszelkich nowych podatków, mówię to wyraźnie, żeby to wybrzmiało, ale skoro mamy maniaków podatkowych w rządzie, bo pan Mateusz Morawiecki zareagował na kryzys, ogłaszając, że na forum unijnym będzie pielgrzymował, żeby wprowadzić trzy nowe podatki, to jest jego ofensywa dyplomatyczna, a na forum wewnętrznym zaproponował, że będzie wprowadzał z zaskoczenia nowy podatek, jak to nazwali, od usług audiowizualnych na żądanie, to może chociaż zrobić to zgodnie z jakąś logiką? Dlaczego nie zabieracie tym, którzy mają najwięcej pieniędzy? Co to za dupochron z przekazywaniem pieniędzy twórcom? Co to za kombinacje? To są wasze „lub czasopisma” Gdyby tu nie było słów „na żądanie”, to największe amerykańskie korporacje by podpadły pod tę ustawę. A tak zrobiliście to w ten sposób, że zapłaci część polskich firm. Suma z tego podatku, z tego, co tu widzę, wyliczenie - kilkanaście milionów złotych. Właśnie sobie wypłacacie z narodowego banku dziesiątki, o ile nie setki miliardów złotych, w ogóle poza kontrolą budżetową, poza kontrolą Sejmu. No co wy wyrabiacie? O co tu chodzi? Kto nam w ogóle to wytłumaczy? Są w tej tarczy też inne ciekawe rzeczy, mogę i o nich powiedzieć kilka słów, chociaż może nie tak zaskakujące, bo są to pomysły Konfederacji, np. zwolnienie z ZUS-u drobnych przedsiębiorców, tych, którzy mają wysoki obrót, nieduży dochód. To myśmy o tym mówili. Zgłaszaliśmy taką poprawkę do pierwszej tarczy, do drugiej tarczy. Proszę bardzo, jest trzecia tarcza, rząd poszedł po rozum do głowy, robi to, co proponowała Konfederacja. Skorzystają na tym ludzie z gastronomii, handlarze, różne niskomarżowe usługi. Okazuje się, że jednak da się zrobić to, co Konfederacja postulowała w wyborach do Sejmu, a więc np. chodzi o elektroniczne doręczenia w sądach. Kto o tym mówił w kampanii wyborczej w zeszłym roku? My - kiedy wyście się bawili w rozgrywki na szczytach hierarchii sędziowskiej. Następna sprawa. Okazuje się, że ZUS nie musi wydawać 25 mln zł po to, żeby rozsyłać wszystkim papierowe informacje o tym, ile mają tzw. składek, które, tak na marginesie, nigdzie się nie odkładają, państwo pewnie doskonale o tym wiecie. Okazało się, że dzięki epidemii można ograniczyć biurokrację w ZUS-ie. Ale mamy też inne ciekawostki, np. kolejne ułatwienia dla imigrantów zarobkowych. W poprzedniej tarczy, pierwszej, drugiej, rząd automatycznie wydłużył pozwolenia na pracę dla imigrantów zarobkowych. Teraz wprowadza dalsze ułatwienia, żeby znieść obowiązek aktualizacji zezwoleń przy zmianie warunków zatrudnienia.

To kwota, o której wy mówiliście, że będzie na koniec roku, a mamy kwiecień. Dziękuję. Zamykam listę osób zapisanych do głosu, do pytań. Informuję, że Prezydium Sejmu na podstawie art. 39 ust. 1 regulaminu Sejmu ustaliło w tym punkcie limit 30 pytań dla klubów według następującego parytetu: Prawo i Sprawiedliwość - 15, Koalicja Obywatelska - dziewięć, Lewica - trzy, Polskie Stronnictwo Ludowe - dwa, a także jedno pytanie dla koła. Jako pierwszy zadaje pytanie pan poseł Andrzej Kosztowniak.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Słyszymy z wypowiedzi opozycji, że nie ma żadnych pieniędzy, nikt niczego nie dostanie, wszystko jest iluzją. Tak trzeba sobie tłumaczyć te wszystkie wypowiedzi. Proszę o informację dotyczącą choćby dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu. Ile przedsiębiorstw z tego może skorzystać, wedle symulacji oczywiście? Z drugiej strony chciałbym, abyśmy dowiedzieli się, ile osób, w symulacjach, może skorzystać choćby ze zwolnienia z opłacenia składek. A trzecią rzeczą jest to, ile osób może również skorzystać z podniesienia kryterium dochodowego do 900 zł w przypadku świadczeń funduszu alimentacyjnego. Pan poseł Dariusz Rosati, klub Koalicji Obywatelskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przedstawiliście projekt tarczy nr 3. Sporo było już mowy na temat tego, co w tej tarczy się znalazło, sporo gorzkich słów pan usłyszał. Chciałem panu zadać pytanie po raz trzeci o to, czego w tej tarczy nie ma. Nie ma w tej tarczy obowiązku testowania pracowników medycznych testami przesiewowymi w sposób cotygodniowy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To już trzeci sezon rządowego serialu pt. tarcza antypracownicza. Mamy już obniżki płac, zapowiedź zwolnień w budżetówce, wydłużenie czasu pracy, a nawet wskazanie przez szefa miejsca skróconego odpoczynku. Zdążyliście zalegalizować obozy pracy w Polsce - brawo. Nie zdążyliście wesprzeć ludzi, którzy tę pracę tracą. Stąd moje pytanie: Czy rząd planuje zostawić ludzi, którzy stracili pracę, zupełnie bez środków do życia? Czy rząd naprawdę sądzi, że te żenujące zasiłki 500 zł, które dostaje i tak bardzo niewiele osób, wystarczą? Otóż nie wystarczą. Jeżeli nie macie swoich pomysłów, skorzystajcie z pomysłów Lewicy. Wprowadźcie natychmiast świadczenie kryzysowe w wysokości 2100 zł na rękę dla wszystkich, którzy stracili źródło utrzymania, bez względu na rodzaj umowy.

Wysoka Izbo! Wszyscy ci, którzy czekali na trzecią wersję tarczy antykryzysowej, naprawdę mieli większe oczekiwania niż to, co zostało tutaj zaproponowane. Tym bardziej te oczekiwania są słuszne, że państwo mieli naprawdę dużo czasu i dużo doświadczeń i wniosków płynących chociażby od rodzimych przedsiębiorców. Dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć: To, co państwo przygotowali, nie przypomina żadnej tarczy 3.0, tylko bardziej przypomina dramat w trzech aktach. Bo czy myślicie, że polski przedsiębiorca, któremu zamknęliście firmę 7 tygodni temu, ucieszy się, że będzie miał szansę złożyć wniosek o dopłatę do odsetek kredytowych? A może ten przedsiębiorca ucieszy się z tego, że są zmienione przepisy o Instytucie Solidarności i Męstwa? Szanowni państwo, naprawdę takich przepisów nam nie potrzeba. Potrzeba życiowych przepisów, które wnoszą cokolwiek do funkcjonowania firm w naszym kraju. Jedyny postęp, jaki widzę, to postęp w liczbie stron tych ustaw. Pierwsza miała 25, druga - 45, ta ma 65% przepisów bardziej skomplikowanych, bardziej niejasnych i nieżyciowych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych pół godziny po zakończeniu pierwszego czytania projektu ustawy z druków nr 344 i 344-A. Bardzo dziękuję. Wracamy do pytań. Kolejne pytanie, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacji.

Mogę mówić? Dziękuję. Panie Marszałku! Przecież nie ma żadnej epidemii, jest to fakt dziennikarski. Takich epidemii mamy kilka rocznie. A wy zabieracie pieniądze z onkologii i dajecie na koronawirusa. Straszycie ludzi i bierzecie ludzi pod but. Już byłoby dawno po epidemii, zmarłoby nie 500 osób, a 3 albo 4 tys. ludzi, ale już byłoby po epidemii. Umrze w końcu 6 tys. osób albo więcej (Dzwonek), ale rocznie gospodarka, dziennie gospodarka traci na tym kilkanaście miliardów złotych. To nie koronawirus jest winien, tylko wy. Pani poseł Barbara Nowacka, klub Koalicji Obywatelskiej.

Panie Ministrze! Tyle dobrych słów, będzie trzecia tarcza, przedsiębiorcy czekają, ludzie pracy czekają. Na razie udało wam się przestraszyć pracowników i oczekują dzisiaj od pana ministra i od pana premiera jasnej deklaracji, że ani w tej, ani w kolejnych waszych pseudotarczach nie będzie mowy o zwalnianiu e-mailem, o zabranianiu ludziom dorabiania, o zwalnianiu ludzi starszych z pracy. Po prostu oczekujemy jako ludzie, jako obywatelki i obywatele tej jasnej deklaracji, że tych antypracowniczych zapisów ani w tej, ani w kolejnych tarczach nie będzie. Jeżeli chcecie rządzić, rządźcie tak, żeby ludzie nie bali się czegoś więcej niż wirusa. Mówicie, że tyle będziecie pomagać przedsiębiorcom. Mało jest tego. Mówicie, że będziecie pomagać rodzinie, wprowadzacie zmiany dotyczące przepisów alimentacyjnych, ale troszeczkę mało. Dlaczego nie zgodzicie się na to, żeby kierowano zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych (Dzwonek) również drogą elektroniczną?

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Mniej więcej tak to wszystko wygląda i właściwie większej pomocy dla przedsiębiorców w tej tarczy nie widać. Natomiast zwracam uwagę, że jednak na tej sali pada ileś pomysłów zarówno w dyskusji, jak i w formie ustaw. Przypomnę, że Lewica złożyła ustawę dotyczącą ochrony miejsc pracy, Lewica złożyła ustawę o świadczeniu kryzysowym, Lewica złożyła ustawę o pomocy przedsiębiorcom w celu pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania. Moje pytanie jest takie: Czy tymi sprawami również rząd się zajmie?

Pan poseł Jacek Protasiewicz, klub PSL-Kukiz. Panie Ministrze! Zachwalał pan tutaj tak bardzo tarczę 3.0, nowy projekt ustawy złożony przez rząd, wymieniając różne aspekty, w tym nie do końca gospodarcze, ale w ogóle pan nie wspomniał o tym, że przy okazji nowelizuje ona Prawo o prokuraturze. Mówiłem o tym wcześniej. Gdyby to jeszcze chodziło o ten 6-miesięczny okres przesunięcia wyborów ze względów zdrowotnych. Dajecie to prawo prokuratorom, nie dajecie zwykłym Polakom. To wasze skrzywienie. Ale po co zmieniacie strukturę rad prokuratorskich kolegiów, zapewniając miejsca zastępcom prokuratora, czyli funkcyjnym mianowanym przez ministra zdrowia? A ja panu powiem, staropolskie przysłowie mówi: łyżka dziegciu zepsuje beczkę miodu.

Panie Marszałku! Mam pytanie do pana ministra Schreibera. Przy okazji mówienia o tym, co zapisano w zmianach do Prawa telekomunikacyjnego, nie zająknął się pan ani słowem, że najbardziej korzystne będą te zmiany dla organu regulującego usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dla prezesa, bo będzie go o wiele łatwiej powołać - wyeliminowano w tych przepisach, w tym projekcie Senat, który do tej pory musiał się zgodzić na daną kandydaturę - i będzie go trudniej odwołać. A dlaczego będzie go trudniej odwołać? Ponieważ wyrzucono z dotychczasowych przepisów możliwość odwołania prezesa, uwaga, za rażące naruszenie prawa, a także jeśli byłoby wobec niego wydane orzeczenie zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa. I teraz pytanie: Czy ma to związek z tym, że pan prezes odpowiada za regulacje rynku pocztowego, który to rynek ma się zająć organizacją wyborów z rażącym naruszeniem prawa? Czy ma to związek z jakimiś przyszłymi interesami, które już być może gdzieś tam w różnych umysłach są założone, a wiecie, że będą one rażącym naruszeniem prawa?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pierwsza, druga, trzecia tarcza i znowu się nie udało. Połowa artykułów tego projektu nie ma nic wspólnego z epidemią. Znów mamy efekt ministerialnej obiegówki, życzeniowe tutti frutti, o nasiennictwie, związku łowieckim, a żeby była odmiana, tym razem, zamiast stawiać maszty, rząd chce łupić takie platformy jak Netflix, choć czasami są one, tak jak w tej chwili, jedynym oknem na kulturę. A jeżeli już jesteśmy przy kulturze, zadam pytanie wicepremierowi Glińskiemu. Czemu znowu nie zadbał o animatorów kultury, którym w tej chwili samorządy na potęgę odwołują konkursy? Nie dostaną zasiłku dla bezrobotnych, opiekuńczego, postojowego, dosłownie nic. Proszę o odpowiedź na piśmie w terminie krótszym niż 77 dni, bo tyle pan wicepremier zwykł trzymać moje interpelacje w szufladzie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejny numer tarczy i kolejne zawiedzione nadzieje przedsiębiorców i pracowników. Za chwilę będziemy mieli więcej numerów tarcz niż wersji Windowsa czy modeli iPhone’a na rynku, a dalej nie będzie rozwiązany żaden problem polskiej gospodarki. Kiedy będzie realna pomoc dla pracowników i firm? Nie pytam, kiedy będą mogli złożyć wnioski, tylko kiedy dostaną pieniądze, kiedy będzie realna pomoc, kiedy na ich konta wpłyną środki na utrzymanie miejsc pracy, na utrzymanie płynności, żeby mogli przetrwać ten trudny okres. Jeśli nadal będziecie tak picować i będziecie taką propagandę uprawiać, to jeszcze wiele, wiele miesięcy firmy będą czekały na pieniądze.

Problem w tym, że we wrześniu może być tak, że już nie będzie miał kto z tej pomocy skorzystać, nie będzie firm, a pracownicy staną się bezrobotnymi.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Trzy podejścia, to trzecie podejście, a tarcza ciągle jak sito. Firmy funkcjonujące w specjalnych strefach ekonomicznych korzystają z ulgi w podatku dochodowym, ale warunek, aby z tej ulgi korzystać, to zainwestowanie określonej kwoty, ale też zatrudnienie określonej liczby osób. Dzisiaj, przy spadku zamówień, przy bardzo istotnym spadku sprzedaży, w wielu przypadkach nie są one w stanie utrzymać zatrudnienia na poziomie określonym w umowie, a niewywiązanie się z tej umowy grozi zwrotem udzielonej pomocy publicznej.

Pani poseł Katarzyna Lubnauer, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie i Panowie Posłowie! Wydawało się, że kolejne tarcze mają służyć temu, żebyśmy my jako Polska i Polacy wyszli z tarczą, a nie na tarczy z tego wyzwania, jakim jest epidemia, natomiast okazuje się, że tarcza najbardziej uderza w kolejne grupy społeczne, tym razem w nauczycieli. Nie wiem, jak - chciałabym o to spytać rząd - w jaki sposób ma pomóc w organizacji pracy szkoły to, że daje się ministrowi prawo do wyłączania zapisów Karty Nauczyciela.

Działacie chaotycznie, działacie wbrew obywatelom, działacie w ten sposób, że mało co idzie na rzeczywiste utrzymanie miejsc pracy. Proponowaliśmy konkretne rozwiązania, np. żeby pozwolić przedsiębiorcom zachować ich VAT, żeby wyłączyć split payment na pewien czas - nie wprowadziliście tego. Proponowaliśmy zwolnienie z ZUS dla wszystkich - nie wprowadziliście tego. Natomiast uderzacie w kolejną grupę społeczną.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przy tarczy 2 większość parlamentarna poparła kilka bardzo dobrych poprawek, które złożyliśmy jako klub Koalicji Obywatelskiej. Nasze poprawki dotyczyły m.in. wydłużenia okresu ważności legitymacji dla studentów i doktorantów, ale również wydłużenia okresu zawieszenia spłat kredytów studenckich do 6 miesięcy. W przedstawionej nowelizacji państwo te poprawki utrzymują. To dobry krok. Ale przypominam, że w chwili gdy procedowaliśmy tarczę 2, Ministerstwo Zdrowia informowało, że szczyt epidemii przypadnie na koniec kwietnia. Tymczasem dziś pojawiają się głosy, że szczyt zachorowań może wystąpić na jesieni. Stąd moje pytanie: Jeżeli szczyt zachorowań faktycznie przypadnie jesienią, to czy zgodzicie się państwo, aby pozytywnie zaopiniować naszą kolejną poprawkę wydłużającą możliwość zawieszenia spłat kredytów na kolejne 3–6 miesięcy? Dziękuję bardzo. Pan poseł Marcin Kierwiński, klub Koalicji Obywatelskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Znowu wielkie liczby, znowu wielkie słowa, tylko bardzo małe efekty tego, co zostało uchwalone wcześniej. Znowu za chwilę dowiemy się od pana premiera Morawieckiego, jak wiele wniosków zostało złożonych, jak wy dzielnie pomagacie, tylko polskie firmy, polscy pracownicy, polscy przedsiębiorcy chcieliby dowiedzieć się, ile pieniędzy już wypłaciliście, ilu firmom pomogliście, ile wniosków rozpatrzyliście, bo o tym ciągle nie mówicie. Proponuję wam, abyście zmienili tę nieustannie powtarzaną frazę: będziemy pomagać na słowo: pomagamy, bo na razie nie pomagacie. Na razie są takie sytuacje, że na 400 wniosków w jednej miejscowości wszystkie są odrzucane. Wczoraj widziałem się z przedsiębiorcami z Ursynowa. Żaden wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Czas przestać mówić, ile jest wniosków. Panie Marszałku! Państwo się chwaliliście, że daliście płynność bankom. Przykład? Kto może w Polsce wziąć kredyt hipoteczny z wkładem własnym 40%? To jest odmrażanie gospodarki?

Gdzie pan się obciął? Wszyscy Polacy chodzą do podziemia fryzjerskiego, kosmetycznego. Czy to jest bezpieczne, że wszyscy się obcinają gdzieś u kogoś w mieszkaniu? Nie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować za debatę, choć muszę powiedzieć, że odbyła się ona w dość specyficznych warunkach. Najpierw zacznę od tych uwag ogólnych. Tarcza.

Jeżeli państwo sami dla siebie używacie takich określeń, to rozumiem, że te żarty są kierowane pod własnym adresem. Cały czas mówiłem, cały czas mówię: to jest rozszerzanie tarczy antykryzysowej, która została zapowiedziana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Było na koniec pytanie, zdaje się, pana posła szanownego. To chciałbym odpowiedzieć: oprócz tego, że 2400 tys. takich wniosków zostało złożonych do wczoraj. Pożyczek łącznie przyznanych, wniosków rozpatrzonych pozytywnie jest 131 tys. Tylko pamiętajmy jedno: powiatowe urzędy pracy są w rękach samorządów.

Idziemy dalej. Ochrona miejsc pracy. Sama liczba wniosków.

Chciałbym tylko państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której też już mówiłem: teraz tym głównym, wielkim instrumentem jest przecież tarcza finansowa. To przygotowana i zapowiedziana przez pana premiera olbrzymia operacja, która została wykonana. Tak jak od początku było zapowiadane, chcemy zrobić wszystko, aby w ostatnich dniach kwietnia, żeby chociaż w ostatnim dniu kwietnia zostało to uruchomione.

75% umarzalnej pożyczki bądź subwencji połączone - o to dopominali się posłowie Lewicy - właśnie, z czym? Z tym, żeby chronić miejsca pracy. Szanowni państwo, przez pierwszy rok nikt nie zapłaci nic - 25% jest umorzone.

Z chwilą, gdy przedsiębiorca zawiera. A więc aż 75% będzie mogło być umorzone, a 50% tej pożyczki będzie mogło być umorzone dzięki utrzymaniu miejsc pracy. Tak samo w sektorze MŚP. Tutaj to będzie 25%, zależne od utrzymania miejsc pracy, ale kwoty są znacznie większe.

36 tys. zł razy ilość pracowników.

Szanowni Państwo! Mówicie o prawie pracy, mówicie o artykułach prasowych, do których się odnosicie, i twierdzicie, że coś jest. Macie projekt ustawy, w którym nie ma takich zapisów. Macie jasną deklarację. Mogę ją złożyć jeszcze raz.

Wręcz przeciwnie, chcemy raczej ratować miejsca pracy.

Chciałbym państwu o czymś powiedzieć.

Jak będzie konieczność, to i częściej.

Zachęcam do pracy w komisjach i do poparcia tego projektu.

Ja przypomnę, że państwo robiliście jedną taką operację, tylko raczej chodziło o to, żeby zabrać Polakom środki z OFE i przekazać je do ZUS-u. Pani marszałek nie potrafiła powiedzieć nawet jako rzecznik rządu, jak to się stało.

Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zawarty w drukach nr 344 i 344-A, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Poproszę panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej panią Marlenę Maląg o przedstawienie informacji. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Parlamentarzyści!

Według posiadanych danych rocznie ponad 115 tys. polskich pracowników przygranicznych pracuje za granicą, przede wszystkim w firmach z siedzibą w Niemczech oraz Czechach.

Od momentu wprowadzenia w Polsce restrykcji w przekraczaniu granicy w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego pojawiły się również ograniczenia dla pracowników przygranicznych, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, ale codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu dojeżdżają do pracy do sąsiedniego kraju. Obowiązek 14-dniowej kwarantanny z jednej strony ogranicza rozprzestrzenianie się COVID-19, z drugiej powoduje ograniczenie w wykonywaniu pracy zawodowej przez Polaków dojeżdżających do pracy za granicą. Co istotne, instytucja obowiązkowej kwarantanny służy nadrzędnemu celowi, jakim jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii i ochrona życia i zdrowia ludzkiego. W ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 polski rząd za pośrednictwem podległych instytucji i służb na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na terenie kraju. Wdrożone obecnie rozwiązania uwzględniają również dane dotyczące zakażeń wirusem w innych państwach, w szczególności tych sąsiadujących z Polską. Zgodnie z przyjętymi zasadami systematycznie przeprowadzana jest ewaluacja zmian, jakie zachodzą w celu realizacji zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Dlatego też dalsze decyzje dotyczące obostrzeń i nakazów zależeć będą od przyrostu liczby zachorowań, wydajności służby zdrowia oraz realizacji wytycznych sanitarnych przez odpowiednie podmioty. Na tym etapie walki z pandemią Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokładają wszelkich starań, aby wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wymiana informacji z instytucjami zagranicznymi uprawnionymi do wypłaty tych świadczeń przebiegały bez utrudnień. Sytuacja pracowników przygranicznych i transgranicznych poddanych kwarantannie w zakresie prawa do świadczeń społecznych z tego tytułu regulowana jest zarówno przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej. Osoby podlegające ustawodawstwu państwa innego niż Polska, ale mieszkające w Polsce, nabywają prawo do świadczeń społecznych z tytułu kwarantanny na podstawie ustawodawstwa państwa, w którym są ubezpieczone. Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji zabezpieczeń społecznych polscy pracownicy przygraniczni w przypadku utraty pracy mogą się rejestrować jako osoby bezrobotne i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych [[Oklaski]] w państwie swojego zamieszkania, a więc w Polsce, pomimo że wszystkie składniki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia na wypadek bezrobocia były za nich opłacane w państwie zatrudnienia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli pracownik przygraniczny zdecyduje się na tymczasową, trwającą dłużej niż tydzień zmianę miejsca zamieszkania: z Polski na państwo zatrudnienia, utraci on status pracownika przygranicznego w rozumieniu unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jaka jest konsekwencja?

W tym celu zwróciliśmy się zarówno do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu rozwiązania problemów pojawiających się w związku z ograniczeniem możliwości (Dzwonek) przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej oraz wykonywania pracy i działalności gospodarczej. W odniesieniu do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek w innych państwach Unii Europejskiej czy obszarów gospodarczych Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii wypracowaliśmy następujące rozwiązania.

Osoba nadal będzie upoważniona do podlegania ustawodawstwu państwa zatrudniającego. W odniesieniu do art. 12 tegoż rozporządzenia, dotyczącego pracowników delegowanych, w przypadku przekraczania maksymalnego okresu delegowania, w trakcie którego możliwe było świadczenie pracy w Polsce, przez pracownika delegowanego do Polski ze względu na COVID-19 polskie instytucje ubezpieczenia na wniosek zagranicznych instytucji będą wyrażały zgodę na wydłużenie okresu delegowania w drodze porozumienia wyjątkowego, co w tej sytuacji właśnie ma miejsce. W przypadku osób wykonujących pracę równocześnie w dwóch lub więcej państwach członkowskich zmiana harmonogramu pracy, w tym powierzenie wykonywania pracy zdalnej i telepracy w państwie zamieszkania lub w innym państwie członkowskim, nie będzie powodować zmiany wcześniej ustalonego obowiązku ustawodawczego.

Wyczerpała pani czas. Dziękuję bardzo. Ostatecznie właśnie decyzje, które są podejmowane, są rozpatrywane w zespole zarządzania kryzysowego. Wnioski są również zebrane z państw ościennych. W przyszłym tygodniu w ramach odmrażania gospodarki zostaną przedstawione.

Jako pierwsza w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pani poseł Teresa Wargocka. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec Informacji Rządu na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Polski oraz poza jej granicami. Szanowni Posłowie! Jeszcze pół roku temu nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, z jakim ogromnym problemem zdrowotnym, społecznym i gospodarczym będziemy musieli się zmierzyć jako klasa polityczna, jaką próbę solidarności i samoograniczenia będzie musiało przejść nasze społeczeństwo. Nowy koronawirus SARS-CoV-2, wywołana nim choroba to bardzo groźny przeciwnik. Choroba, która stała się światową pandemią, zburzyła spokój społeczny, zatrzęsła światową gospodarką. Rząd, podległe mu służby, spółki Skarbu Państwa, samorządy, wolontariusze, wszyscy ludzie wielkiego serca w miarę swoich obowiązków, kompetencji podjęli stosowne działania. Dzisiaj, po 2 miesiącach od pierwszego zachorowania należy stwierdzić, że udało nam się zapanować nad rozprzestrzenianiem się choroby. Utrzymujemy spłaszczoną liczbę wzrostu zachorowań, a ilość zakażeń i zgonów jest najniższa w Europie. System ochrony zdrowia jest w pełni przygotowany do walki o życie i zdrowie Polaków. Mamy odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej. W tej chwili w naszym kraju działa 20 szpitali jednoimiennych, tj. ponad 10 tys. miejsc, 79 oddziałów zakaźnych, uruchomiliśmy od zera 80 laboratoriów, mamy zapasy testów. Każdy wybiera sobie sposób mówienia taki, jaki uważa. Nie ma problemów ze sprzętem ochrony osobistej, z ilością testów. Polskie społeczeństwo przestrzega zasad izolacji, stosuje się do wprowadzonych obostrzeń i niewątpliwie ma ogromne zasługi w tym, że koronawirus w Polsce jest pod kontrolą. COVID-19 to również ogromny wpływ na gospodarkę. Dlatego rząd przygotował tarczę antykryzysową, tarczę finansową. Elementy tej tarczy są już realizowane, składane są wnioski, wypłacane są pierwsze pieniądze. To jest ok. 15% PKB. Nikt nie mógł takiej epidemii przewidzieć. Obok kosztów zdrowotnych, gospodarczych są również koszty społeczne - i te koszty społeczne głównie przejawiają się lękiem o utrzymanie miejsca pracy i utrzymanie dochodów rodzin. Takie lęki przeżywają w tej chwili miliony polskich pracowników. Dzisiejsza informacja rządu dotyczy wąskiego wycinka tego problemu, związanego z zatrudnieniem transgranicznym. Tak jak pani minister mówiła, ponad 100 tys. polskich pracowników pracuje za granicą w sferze transgranicznej, głównie w Niemczech i w Czechach. Wprowadzona od 27 marca kwarantanna zdecydowanie wpłynęła na trudną sytuację tych pracowników i postawiła ich przed dylematem, czy zamieszkać w kraju zatrudnienia, czy pozostać w Polsce i przebywać z rodziną. Z informacji pani minister wynika, że prace ministerstwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS-u są prowadzone, że sytuacja jest monitorowana, że system zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej jest analizowany. Ministerstwo wprowadziło pakiet rozwiązań dla pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej w oparciu o rozporządzenie o pracownikach delegowanych. Szanowni Państwo! Na pewno problem jest, problem musi być rozwiązany w porozumieniu z innymi agendami unijnymi. Dlatego cztery etapy, które przedstawił pan premier Morawiecki, to są etapy odmrażania polskiej gospodarki. Mam przekonanie, że również pracownicy transgraniczni przyjmą te działania rządu jako pozytywne i przyjmą ten główny kierunek (Dzwonek), tę zasadę, że dalsze znoszenie zakazów musi odbywać się tylko pod rygorem oceny stanu epidemicznego w Polsce i w krajach, z którymi graniczymy. Teraz głos zabierze pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście czas pandemii to czas bardzo trudny, to czas dramatycznych wyzwań, to czas próby i niełatwych decyzji, ale to także czas sprawdzenia, jak działa rząd, jakie decyzje podejmuje, sprawdzian jego odpowiedzialności za losy państwa i obywateli. Jednak jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w naszym kraju, to prawie w większości przypadków Polacy zostali zostawieni sami sobie. I zamiast pomocy dostają coraz dłuższe konferencje prasowe, coraz więcej słów, ale coraz mniej konkretnych informacji. Nawet dzisiejsza informacja pani minister to właściwie dwie informacje: instrukcja, jak zarejestrować się jako bezrobotny, i to, że w przyszłym tygodniu zostanie pokazany jakiś plan. Jakiś plan, a ludzie oczekują konkretnych informacji. W zeszłym tygodniu rozmawiałam z kobietami mieszkającymi w strefie przygranicznej, które opowiedziały swoje historie. Matka samotnie wychowująca dzieci musiała zostać w Niemczech, bo gdyby wróciła do kraju, straciłaby pracę, nie miałaby środków na utrzymanie dzieci. Dzieci muszą być same. W takich sytuacjach ludzie dokonują dramatycznych wyborów. Widzieliśmy protesty, widzieliśmy protesty ludzi, widzieliśmy dramatyczne sceny, dzieci płaczące na widok swoich ojców. Państwo musi podejmować decyzje i musi tym ludziom pomagać. Te osoby, z którymi rozmawiałam, od państwa polskiego nie dostały żadnej pomocy.

Bardzo trudno będzie wrócić i na nowo odzyskiwać klientów, i budować swój potencjał, ale także zasobność naszego kraju. Powinniśmy podjąć decyzje, podać konkretny plan wychodzenia z tego, konkretne daty. Ludzie muszą wiedzieć, czego się mogą spodziewać. Tak, to ma być bezpieczne.

Jeżeli będziemy testować, będziemy mogli szybciej pozwolić ludziom wracać do normalności, ale trzeba odważyć się i podjąć takie decyzje. Mówimy o tym od kilku tygodni. Mam wrażenie, że ci ludzie, którzy stworzyli te wspaniałe euroregiony, coś, o czym marzyliśmy, współpracę pomiędzy krajami tych małych ojczyzn, zostali zostawieni sami sobie. Nawet przedstawiciele krajów, Czech, Niemiec, apelują do polskiego rządu o to, żeby wspólnie wypracować rozwiązania. Rząd milczy i nie pochyla się nad tym. I naprawdę uważam, że dzisiejsza wypowiedź pani minister, w której nie było ani jednego konkretu, ani jednego pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji, świadczy o tym, że wy do tego jesteście w ogóle nieprzygotowani i w ogóle o tym nie myślicie. I gdyby nie protesty ludzi, które były i które mają być 1 maja, i gdyby nie to, że posłowie opozycji ciągle zadają pytania, pytają, co zrobiliście w tej sprawie, to tej informacji by nie było. Tak źle przygotowanej informacji w tym Sejmie jeszcze nie słyszałam. Ale przecież nie chodzi o to, żeby ci ludzie byli bezrobotni, tylko żeby utrzymać ich miejsca pracy i żeby mogli wrócić do normalnego życia. Dlatego w imieniu klubu Koalicja Obywatelska zgłaszam wniosek o odrzucenie informacji rządu. Naprawdę to była bardzo skandaliczna informacja i jest mi po prostu wstyd, że rząd lekceważy Polaków, nie pochyla się nad ich sprawami. I naprawdę możemy codziennie pytać o strefy transgraniczne, możemy pytać o lekarzy, możemy pytać o nauczycieli, o każdy obszar naszego życia. Wy nie robicie nic, tylko mówicie, że przedstawicie plan. Ja bym nawet chciała poprosić o taką informację rządu, o to, żeby rząd przedstawił konkretne osoby, którym pomógł, żebym mogła poznać osoby, które rządowi zawdzięczają pomoc i wiedzą, że mogą wyjść z kryzysu, bo na razie to są tylko obietnice. Słowa, słowa. Pani poseł Katarzyna Kotula, klub Lewicy. Panie Marszałku! Do pana premiera dzisiaj się zwracam jako do osoby decyzyjnej. 4 maja otwiera pan galerie handlowe, hotele, żłobki i przedszkola. A czy wie pan, że 26 kwietnia dzieci w niemieckich powiatach przygranicznych wróciły już do szkoły? Dziś dzieci mieszkające w Polsce, 5 km dalej, nie mogą realizować swojego obowiązku szkolnego. My wiemy, że z pozycji Warszawy to tabele w Excelu i statystyki, ale z pozycji pogranicza to konkretni ludzie i konkretne historie. To pracownicy służby zdrowia, mediów, urzędów, szkół, lokalnych firm małego i średniego biznesu. To pani Ola, która samotnie wychowuje dwójkę dzieci i mieszka po niemieckiej stronie, ale w Polsce ma swoją firmę, do której nie może teraz dojechać. Ale też pani Monika, mieszkająca po polskiej stronie nauczycielka, która nie może wrócić do pracy w szkole po niemieckiej stronie, choć dojazd samochodem zajmuje jej tylko 10 minut. Wielu Polaków straciło pracę nie dlatego, że nie mogą pracować, tylko dlatego, że pan im to uniemożliwił. To ok. 250 tys. polskich obywateli. Ale łącznie kryzys ten dotyczy miliona osób, bo ludzie ci mają rodziny i dzieci. Osób, które zostały bez pracy. To Polacy zatrudnieni w hucie w Trzyńcu, kopalni w Karwinie czy centrum medycznym w Hawierzowie, gdzie produkuje się artykuły medyczne, z których korzysta także Polska. Niejednokrotnie ci, którzy zdecydowali się na pozostanie w Czechach czy w Niemczech, aby móc pracować, zarabiać na chleb, na życie, na rodzinę, legalnie, nie mogą widywać się ze swoimi bliskimi, którzy mieszkają czasami tylko kilka kilometrów dalej, często po drugiej stronie jednego mostu. W czasie piątkowych protestów widzieliśmy rozdzielone rodziny, stały czasami 2, 3 m od siebie, oddzielone ogrodzeniem i wojskiem z bronią. Tymczasem mieszkaniec Łodzi pokonuje większą odległość i zupełnie legalnie może codziennie dojeżdżać do pracy, np. w Warszawie. Panie premierze, regularnie chwali się pan, jak to bardzo Polska przoduje w dobrych rozwiązaniach, a przecież koronawirus nie ma narodowości, nie zna granic. Warto zaznaczyć, warto pokazać, jakie są statystyki. Jeśli chodzi o koronawirusa, przykład: duży powiat Uckermark, który ma ponad 120 tys. mieszkańców, to na dzień dzisiejszy tylko 10 zachorowań, podczas gdy graniczący z nim powiat gryfiński z 82 tys. ludności to 31 zachorowań. Okręg Löcknitz-Penkun to jeden przypadek zachorowania, a graniczący z nim teren Szczecina to 46 przypadków. Panie premierze, ci obywatele są Polakami, ten rząd to także ich rząd, a pan jest ich premierem. Tymczasem to rządy landów Brandenburgii czy Meklemburgii bardziej troszczą się o Polaków niż ich własne państwo. Zarówno polska, jak i niemiecka czy też czeska strona apelują do rządu, aby otworzyć mały ruch graniczny, utworzyć jakiekolwiek rozwiązania.

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sytuację w kraju należy oceniać z różnych stron, a gdy chodzi o dramaty ludzkie, należy rozpatrywać z każdej możliwej do przewidzenia strony. Patrzymy nie tylko przez pryzmat kawalera z wysoką emeryturą i całkiem niezłym uposażeniem czy bankiera, który, choć miał ogromny majątek, dziś udaje, że go nie ma, ale przede wszystkim przez pryzmat dramatów ludzkich. Rząd w swoich decyzjach w zakresie walki ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią pominął wiele grup społecznych, głównie pracowników, którzy w tzw. tarczy antykryzysowej zostali pozostawieni sami sobie. W przeddzień obchodów święta pracy chciałbym przypomnieć wam o dramacie pracowników transgranicznych. To tysiące Polek i Polaków mieszkających na terenach przygranicznych takich jak Zgorzelec, Lubawka, Bogatynia, Zawidów, Porajów, Kamienna Góra czy też cały teren Śląska Cieszyńskiego. Wszyscy oni decyzjami rządu Mateusza Morawieckiego zostali dzisiaj bez pracy i środków do życia. Już teraz mają problemy z opłaceniem bieżących rachunków, a co dopiero z zakupem niezbędnych do życia produktów. Zmuszeni walczyć o swoje miejsca pracy, wyszli na ulicę w wielu miejscowościach w całej Polsce. W ubiegły piątek ogrodziliście ich policją, wojskiem z bronią i nagraliście jak przestępców. Dla was nie liczy się życie ludzi, których wobec władzy uprzedmiotowiliście. Mają być posłuszni, nie protestować i głosować bez żadnego trybu na kandydata, którego im wskażecie. Lewica nie może zgodzić się na takie traktowanie polskich rodzin i patrzeć, jak ignorancja władzy prowadzi do ich zubożenia. Pracownicy transgraniczni powinni być traktowani tak jak zawodowi kierowcy, którzy mogą przekraczać granicę bez żadnych problemów. Żądamy, aby takie same decyzje podjąć wobec pracowników świadczących pracę na terenie Czech czy Niemiec. Przy zabezpieczeniu granic w zaplecze sanitarne na pewno to się uda. W tym trudnym momencie posłowie i posłanki Lewicy. m.in. Robert Obaz, Katarzyna Kotula, byli z pracownikami na granicy. Popieramy ich protest. W imieniu klubu Lewicy wnoszę o odrzucenie informacji rządu na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi pani poseł Jolanta Fedak - zdalnie. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Nie chodzi tylko o Polaków, którzy pracują po drugiej stronie granicy, ale także chodzi o młodzież, która uczy się po drugiej stronie granicy, chodzi też o osoby, które są leczone po drugiej stronie granicy, i odwrotnie. Chciałabym państwa bardzo mocno przekonać do podjęcia decyzji, które są oczekiwane przez mieszkańców dziewięciu województw przygranicznych. Od czasu odbudowania w Polsce samorządu terytorialnego w 1990 r., a szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wzdłuż granic Polski nastąpił bardzo pozytywny proces integracji społeczeństw po obu stronach granicy. Dziś dla wielu Polaków mieszkających z tej strony granicy i dla obywateli Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji z drugiej strony granicy przygraniczne miasta oraz ich infrastruktura, szkoły, szpitale, zakłady pracy, kościoły, targowiska, punkty usługowe stały się po prostu wspólne. Mieszkańcy pogranicza razem z nich korzystają i są bardzo silnie związani codzienną egzystencją. Od wielu lat przekraczają granice po to, żeby korzystać z tych instytucji i placówek, a także firm, bo mają tu po prostu najbliżej i najbezpieczniej. To jest największy motor napędowy rozwoju terenów przygranicznych. Powstało także wiele mieszanych rodzin, chociażby Polacy w coraz większej liczbie zasiedlają osiedla po drugiej stronie granicy.

Tym samym wszystkie obawy dotyczące germanizacji zachodnich terenów Polski, tak często wcześniej zgłaszane, nie mają po prostu racji bytu. To Polacy stali się bardziej dynamiczni, mają dużą siłę przebicia. Coraz częściej Niemcy pracują w Polsce. Wzajemnie korzystamy z transgranicznej oferty oświatowej, zdrowotnej, usługowej. Taki stan rzeczy dotyczy większości naszych granic. Zachodzą niespodziewane zmiany, bo to nie tylko Volkswagen czy BMW inwestują w Polsce, ale także polskie zakłady inwestują po drugiej stronie granicy, w Niemczech. Takim przykładem jest firma córka Azotów Tarnów S.A., która kilometr od Guben wybudowała fabrykę, w której pracują mieszkańcy Gubina.

Mam świadomość powodów, dla których ta granica jest zamknięta, ale przecież mogą ją przekraczać przedstawiciele rożnych służb, np. służb ratowniczych czy Straży Granicznej, służb administracji celnej. A zatem dlaczego nie mogą przekraczać ich sąsiedzi, którzy często obok nich mieszkają i którzy także mają po prostu związane z tym pograniczem swoje życie. Chciałabym także podkreślić, że wielu ludzi korzysta ze szkół i wyższych uczelni po drugiej stronie granicy, bo jest po prostu najbliżej. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś rozpoczął edukację po drugiej stronie granicy, po prostu powinien ją dokończyć. A już w tej chwili szkoły po drugiej stronie granicy są otwierane. Polska przecież szczyci się takimi modelowymi rozwiązaniami miast podzielonych granicą, chociażby Słubice - Frankfurt nad Odrą (Dzwonek), Gubin - Gubin, Zgorzelec - Görlitz, Cieszyn - czeski Cieszyn, gdzie stworzono wspólne systemy komunalne korzystne dla osób z obu stron granicy. Jeszcze raz bardzo proszę, żeby prośbę osób pracujących po drugiej stronie granicy, a mieszkających w Polsce i odwrotnie. Nie ma takiej możliwości, żeby zostawić tych ludzi absolutnie samych i nie robić w tej chwili nic. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu koła Konfederacja głos zabierze pan poseł Krzysztof Tuduj. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Konfederacja apeluje do rządu: otwórzcie granice dla pracowników transgranicznych. Apelujemy dzisiaj, apelowaliśmy wczoraj na konferencji prasowej, apelowaliśmy w zeszły czwartek w Cieszynie na konferencji prasowej. Trzeba zrozumieć sytuację pracowników transgranicznych. To są ludzie, którzy mają nierzadko bardzo małą odległość do pokonania z domu do pracy. To są ludzie, którzy zostali rozdzieleni, rodziny zostały rozdzielone tą przymusową kwarantanną. Zamknięcie granic jest słuszne, ale niezrozumienie sytuacji pracowników transgranicznych jest po prostu wylewaniem dziecka z kąpielą. To jest błąd. Apelujemy: ta sytuacja musi się jak najszybciej skończyć. To jest grupa społeczna, którą rząd pominął. Mało inteligentnie zachował się w stosunku do tej grupy i okaże się, że będą większe skutki zamknięcia granic, niezrozumienia potrzeb pracowników transgranicznych niż samej walki z koronawirusem. Dlatego apeluję z tego miejsca do rządu: natychmiast, jak najszybciej wyjdźcie naprzeciw potrzebom tych ludzi, wyjdźcie naprzeciw potrzebom Polaków, którzy mieszkają przy granicy. Przecież dochodzi już do protestów. Te protesty na pewno nie zwiększą poziomu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o walkę z zarazą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! O kim tutaj mowa? O ludziach wyjątkowych, tak zdeterminowanych, żeby pracować, że szukali tej pracy aż za granicą, aż za cenę rozłąki, chwała Bogu, do tej pory krótszej, nie dłuższej, czasowej z rodziną. I teraz tym ludziom pani minister Maląg proponuje bezrobocie. Ja mam nadzieję, że za sprawą tych protestujących ludzi i za naszą sprawą pani minister Maląg będzie stała szybciej, a nie później wobec takiej perspektywy. Czy poszuka uczciwej pracy, choćby i za granicą, czy też ustawi się w kolejce po zasiłek? To jest świat postawiony na głowie, także ten komunikat, który fałszywie został zatytułowany sprawozdaniem, informacją o tym, jak rząd pracuje nad umożliwieniem. Bo przecież rząd najpierw nie napracował się wiele, bo jednym ruchem uniemożliwił uczciwą pracę setkom tysięcy Polaków wraz z rodzinami.

To jest właśnie perspektywa tej Izby, to jest perspektywa urzędów centralnych. Setki tysięcy uczciwie pracujących ludzi to jest wąski margines. Nie, marginesem społecznym jesteście wy, którzyście nigdy inaczej nie pracowali, jak tylko na etacie państwowym, którzyście nigdy nie szukali uczciwej pracy, ponieważ. Pani marszałek też się zgłasza rozumiem do tej kategorii, tak? Pani marszałek po raz kolejny będzie próbowała recenzować moje wystąpienie a vista. Szanowni Państwo! Koło Konfederacja apeluje ustami pana posła Tuduja, ustami naszego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztofa Bosaka, uparcie powtarzamy: wypuście naród z kwarantanny. No przecież jeżdżą - chwała Bogu, z lękiem to powiem, bo może coś wymyślicie, żeby im przeszkodzić - kierowcy tirów przez granice i nie siedzą 2 tygodnie w kwarantannie.

Rzecz jasna, wzywamy do tego, żeby ogół Polaków został z kwarantanny wypuszczony, i wnioskujemy o odrzucenie tego pseudoraportu. Dziękuję za uwagę. Jeszcze będą pytania, pani poseł.

Proszę nie przypisywać mojej osobie lekceważenia jakiejkolwiek grupy społecznej, jakiegokolwiek problemu, jaki mają ludzie. Nie jestem takim człowiekiem, nie jestem takim politykiem.

W tym fragmencie, który wypowiedziałam, było pokazane tło: lęk społeczny przed bezrobociem i brakiem środków utrzymania. 14 mln polskich pracowników zatrudnionych w Polsce również przeżywa te lęki, bo nie wiemy, czy koronawirus będzie trwał miesiąc, dwa miesiące, pół roku czy rok.

Tak.

Pani reprezentuje zły reżim, zły rząd. I z tego powodu do pani adresowałem moje wystąpienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska. Lista nie była w żaden sposób ograniczona. Dziękuję bardzo. Dobrze, pani marszałek, dziękuję. Słowa, które tu dzisiaj padły, to jest w ogóle. Pani mówiła kompletnie nie na temat, kompletnie nie na temat. Tu chodzi o ludzi, którzy mają firmy usługowe, które świadczą usługi Polakom, Niemcom, Czechom. Stawiam tezę: wy zlikwidowaliście ruch przygraniczny, bo wam potrzebne to było do tego, żeby pan Morawiecki mógł mówić, że Unia Europejska nie działa. Z powodów ideologicznych zamknęliście, żeby mówić: Unia nie działa, zobaczcie. Dlatego zamknęliście granice, dlatego to wszystko stworzyliście. Niech pan lewobrzeżną Warszawę oddzieli od prawobrzeżnej, jest rzeka, są mosty, i niech pan powie: Ludzie, żyjcie, będzie mniej koronawirusa.

Dlaczego? Bo oni badają. Stworzyli system, dogadali się, badają ludzi przekraczających granicę. Kiedy pan Morawiecki i pan Duda byli na granicy u tych ludzi (Dzwonek), u tych zdesperowanych ludzi, którzy walczą o swoje miejsca pracy? Kiedy pan Duda i pan Morawiecki u nich byli? To jest pogarda, co zaproponowaliście z tymi zasiłkami dla bezrobotnych, pani minister. Bardzo proszę, żebyśmy stosowali zasady. Ja poprzedzam pana nazwisko sformułowaniem: pan poseł, a więc bardzo proszę: pan premier Morawiecki, pan prezydent Andrzej Duda. Bardzo proszę, pani poseł. Zajęci usługą pocztową pseudowyborów nadal nie dostrzegacie, pani minister, zapaści pracy na pograniczu. Nie słyszycie głosów tysięcy Polaków, którzy zostali bez pracy i bez możliwości zarobkowania. 15 marca zamknęliście granice i zostawiliście ludzi samych sobie, z problemami, z dylematami i bez pieniędzy, i udajecie, że to nie jest wasz problem. Ludzie protestują na granicach. Piszą do rządu petycje. Apelują do was samorządy i apelują do was euroregiony. W Kudowie, w Cieszynie, w Zgorzelcu, w Kołbaskowie na granicy nadal jest paraliż i zaczynają się ludzkie dramaty. Dziś jest 29 kwietnia, a minister pracy w rządzie Mateusza Morawieckiego mówi do was: Drodzy pracownicy transgraniczni, możecie rejestrować się jako bezrobotni albo możecie wykonywać telepracę.

Pytanie zada pan poseł Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Zamknęliście granice. Wiele osób ma szlaban, ale to nie jest szlaban tylko na przejazd. Dla wielu z nich to szlaban na pracę, szlaban na możliwość zarabiania pieniędzy i często szlaban na kontakt z rodziną. Symbolem rozpaczy tych ludzi stał się mały chłopiec, który na granicy przytulał swojego tatę przez metalowy płot. Przestańcie udawać, że tego problemu nie widzicie. Tylko u nas, w województwie zachodniopomorskim, ten problem dotyczy 20 tys. Polaków, którzy codziennie przekraczali granicę, jadąc od pracy. Waszą rolą i obowiązkiem jest udzielanie im pomocy, więc zamiast wysyłać ich na przymusową kwarantannę, wyślijcie im specjalne przepustki. Otwórzcie dodatkowe przejścia graniczne, gdzie będą kontrole sanitarne i dodatkowe testy. To są te sprawy, na które dziś ci ludzie czekają, więc zamiast zajmować się organizacją wyborów, zajmijcie się [[Dzwonek]] udzielaniem pomocy tym ludziom. Pytanie zada pan poseł Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Problem współpracy transgranicznej jest niezwykle ważny i istotny. Ale to jest także powodem tego, iż te relacje i związki pomiędzy wspólnotami po obu stronach granicy: polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko-litewskiej czy polsko-słowackiej są stosunkowo mocne. Relacje dotyczą nie tylko kooperacji podmiotów gospodarczych, nie tylko edukacji, służby zdrowia, ale także wielu ważnych spraw międzyludzkich.

Pani Minister! Niewybaczalne i nieakceptowalne jest to, że pani resort nie przygotował (Dzwonek) takich przepisów prawa, które umożliwiałyby podejmowanie właśnie tych relacji, przede wszystkim działalności gospodarczej, ale także zapobiegałyby wielu ludzkim dramatom. Pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ponad 12 lat temu na granicznych drogach i szlakach przecięliśmy szlabany i połączyliśmy ludzi. Historyczne krainy, takie jak np. Orawa, Spisz czy Śląsk Cieszyński, przestały traktować granicę jako cokolwiek. Dla nich granica stała się miejscem do współpracy, do robienia wspólnych biznesów. Myśleliśmy, że ten czas przywrócenia szlabanów na granicę już nigdy nie nastąpi. Niestety PiS postawił na nowo szlabany, brutalnie rozdzielił rodziny, często ludzie musieli decydować o tragicznych wyborach: czy zostać w domu, czy kontynuować swoją pracę za granicą. Zlikwidowaliście setki czy nawet tysiące rodzinnych firm, które z tego żyły. Dzisiaj na targowisku w Jabłonce czy w Nowym Targu przedsiębiorcy mówią: granice zamknięte, Słowaków nie ma, z czego mamy żyć? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przychodzimy dzisiaj z dramatycznym apelem setek tysięcy polskich rodzin rozdzielonych murem, który budujecie, nie pozwalając na możliwość pracy tym, którzy często do pracy mają 5 czy 6 km, tak jak mieszkańcy Lubawki. 1 tys. pracowników powiatu kamiennogórskiego nie ma pracy, nie ma możliwości przejechania do pracy, czeka ich za chwilę zwolnienie, tak samo jak 20 tys. Dolnoślązaków przejeżdżających codziennie przez granicę w Zgorzelcu i Görlitz. Dzielicie Polaków. Część osób zmuszona jest do tego, żeby ze swoimi dziećmi mieszkać w hotelach, prowadząc telepracę z hoteli niemieckich, bo obawiają się, że stracą pracę. Chodzi o polskie firmy, które zdobywały przez lata niemieckie i czeskie rynki zbytu, a dzisiaj tak naprawdę tracą te rynki, po prostu plajtują. Dlaczego pięciu uczniów, maturzystów z Polic może bez kwarantanny przekraczać granicę, bo tam kończą matury, a młodzież z Görlitz (Dzwonek) nie może tego zrobić? Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska.

Pani Minister! Wysoka Izbo! W tych dniach na granicach, także w naszym Cieszynie, protestują zdesperowani ludzie. Jeszcze kilka tygodni temu kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, powiatu bielskiego, żywieckiego, Bielska-Białej wyjeżdżało do pracy, by prowadzić biznes w Czechach czy na Słowacji. Nie mogli znaleźć pracy w Polsce, wzięli sprawy w swoje ręce, podjęli pracę, tam prowadzą biznes. Należy im się szacunek, pani minister. Rząd PiS nieprzemyślanym zamknięciem granic i tą obowiązkową kwarantanną pozbawił ich środków do życia, nic w zamian nie proponując, okazując brak szacunku, rozdzielając rodziny. PiS nie rozumie, że w takich miejscach jak Śląsk Cieszyński nawet 30% mieszkańców jest zależnych od dochodów właśnie za granicą. Rząd Republiki Czeskiej to rozumie i tam nie wprowadzono takich ograniczeń. Dziś, szanowna pani minister (Dzwonek), czas proszenia się skończył.

A jeżeli państwo tego nie rozumiecie, to zapraszamy do nas, do Cieszyna. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mieszkam na południe od Raciborza. Kilkaset metrów za moim domem jest czeska fabryka, w której pracuje kilkuset moich sąsiadów, a w całym Moravskoslezskym kraju, czyli odpowiedniku województwa śląskiego, pracuje 12 tys. Polek i Polaków.

Jednocześnie przez te przejścia mogą przejeżdżać rolnicy, którzy uprawiają pola po obydwu stronach granicy. Jaka jest różnica?

Można znaleźć racjonalne rozwiązania, dedykowane przejścia graniczne małego ruchu tylko dla tych pracowników, którzy i tak są badani w swoich zakładach pracy.

Panie Premierze! Bardzo proszę. Panie Pośle Kaczyński! Wysoka Izbo! W związku z licznymi apelami moich wyborców zamieszkujących tereny przygraniczne, by pozwolić im pracować za granicą, zwracam się do państwa z pytaniem: Dlaczego tym nielicznym Polakom, którzy jeszcze nie stracili pracy, bo inne kraje dbają o nich bardziej niż ich własne państwo, uniemożliwiacie tę pracę? Jest to być może już jedna z ostatnich grup społecznych, które nie czekają na skąpą, a najczęściej iluzoryczną pomoc ze strony rządu, tylko chcą, by pozwolić im pracować, by tylko państwo nie przeszkadzało, by pozwoliło pracować, zarobić na życie swoje i swoich rodzin. Dlaczego wasze chore fobie, wasz strach przed zagranicą chcecie przerzucać na lokalne społeczności, które żyją w dobrych relacjach, które czerpią to, co najlepsze z obu stron granic? Nie mierzcie wszystkich swoją miarą.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Posłowie i posłanki Lewicy już takie konkretne propozycje składali, chociażby Przemysław Koperski, poseł Lewicy, składał taką interpelację do pana ministra Jacka Sasina, by otworzyć więcej przejść granicznych, koleżanka Anita Kucharska-Dziedzic osobiście musiała interweniować w sprawie tzw. zbiorowej kwarantanny, w przypadku której warunków zupełnie nie było. Czyli tak naprawdę chodzi o to, co państwo robicie, z jednej strony zamykacie granice, nie korzystacie z pomysłów, które już padają, a z drugiej strony posłanki i posłowie Lewicy muszą interweniować na granicy, tak jak koleżanka Kotula, tak jak poseł Obaz (Dzwonek), by wiedzieć, co mają z tym zrobić. Więc ja proponuję, żebyście państwo czerpali z tych doświadczeń, które my tutaj mamy, i monitorowali to, co robią wojewodowie, bo akurat w województwie lubuskim są skandaliczne warunki, jeżeli chodzi o tzw. kwarantannę zbiorową. Pan poseł Krzysztof Śmiszek, Lewica. Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać w imieniu setek tysięcy Polek i Polaków, którzy mieszkają i pracują w strefach przygranicznych, o to, czym kierował się rząd, narzucając takie barbarzyńskie kryteria nakładania kwarantanny na tych mieszkańców. Proszę mi powiedzieć, ale także proszę powiedzieć tym setkom tysięcy naszych rodaków, jak to jest, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w transporcie międzynarodowym z tej kwarantanny są zwolnieni, a fryzjerka, lekarz czy budowlaniec, który pracuje 3, 5, 7, 15 km od polskiej granicy po stronie niemieckiej czy czeskiej, jest taką kwarantanną objęty. Jak to jest, że kierowca ciężarówki może przejechać całą Europę, a fryzjerka ze Zgorzelca tej granicy przekroczyć nie może? Dlaczego stawiacie ludzi przed dramatycznymi wyborami: albo bezrobocie i bieda, i brak pieniędzy na życie, albo rozłąka z rodziną i dramaty ludzkie? Gdzie jest w tym wszystkim logika? Gdzie jest jakaś empatia i gdzie jest współczucie? Gdzie jest jakiś konkretny plan? Fundujecie naszym rodakom piekielny wybór pomiędzy rozpaczą a biedą. Wsłuchajcie się wreszcie w głosy samorządowców z Lubawki, Szczecina, Zgorzelca i Cieszyna i ich odpowiedników z drugiej strony granicy. Oni mają odpowiedzi, oni mają pomysły, jak te dramaty rozwiązać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! To, co dziś dzieje się na granicach, to jest nie tylko problem tych ludzi, którzy tam mieszkają, to jest nasz problem, wszystkich, bo niedopuszczalne jest, żeby po ponad 20 latach od otwarcia niektórych granic i kilkunastu lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej mierzyć się z takimi wielkimi dylematami jak ten, czy ktoś, jak przekroczył niechcący granicę, nie będzie mógł za chwilę wjechać do Polski, bo pomylił się i przejechał gdzieś na jakimś rozdrożu przez granicę na 5 minut.

Bo to dzisiaj samorządowcy odpowiadają na te wszystkie pytania i brak im pomocy, brak im słów, brak im wsparcia, które rząd [[Dzwonek]] powinien zafundować nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyznam się szczerze, że jak wysłuchałem tej informacji, to jednej rzeczy jestem pewny: wy nas tutaj z tej centralnej Polski kompletnie nie rozumiecie, nie wiecie, co my tam czujemy w tych rejonach nadgranicznych - ja akurat jestem ze Szczecina. Nic w tej informacji takiego nie ma. Przecież to jest prosta sprawa - zbadać ilość zakażeń w promieniu 30 km po jednej i po drugiej stronie granicy i powiedzieć: rzeczywiście jest poważny problem, nie możemy otwierać tych granic, albo powiedzieć: rzeczywiście 30 km w tę i w tę stronę możemy granicę przekraczać. Ja apeluję: zróbcie państwo taką analizę i po prostu powiedzcie uczciwie, że można coś takiego zrobić. Bo ja w to głęboko wierzę i widzę, że można to zrobić. Jest stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące tego, że powinniśmy otworzyć granice. Pytanie: Jak Polska, jak polski rząd [[Dzwonek]] do tego podchodzą i co planujecie w najbliższym czasie w tym zakresie? Pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Pani Minister! Ja w zeszłym tygodniu byłem w Cieszynie, po to żeby wesprzeć pracowników transgranicznych i lokalnych działaczy, którzy się za nimi ujmują w sprawie możliwości legalnego zarobkowania, normalnego życia. W tej chwili ci ludzie, którzy protestowali w ostatnich dniach w Szczecinie, w Zgorzelcu, w Cieszynie, w innych miastach przygranicznych, są postawieni przed dramatycznymi wyborami: albo oderwać się od rodziny i zarabiać na życie, albo zostać z rodziną i stracić źródło utrzymania. W takiej sytuacji polski rząd nie powinien tych ludzi stawiać. Czym innym jest ruch transgraniczny, ruch turystyczny, ruch międzypaństwowy, okazjonalny, a czym innym jest przemieszczanie się czy to nas mieszkających tuż pod Warszawą do pracy w centrum Warszawy, czy tych ludzi o kilkadziesiąt kilometrów do swojego miejsca pracy. Pozwólmy tym ludziom normalnie pracować. Otwórzmy gospodarkę. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Pierwsze pytanie: Dlaczego działacie wbrew wytycznym Komisji Europejskiej? Pani minister dokładnie wie, że 30 marca Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie swobody przepływu pracowników podczas epidemii. Komisja Europejska zaleca, żeby pracownicy z obszarów transgranicznych mogli swobodnie przemieszczać się do swojej pracy, utrzymać źródła utrzymania. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, pani minister, to testy. Nie wiem, czy pani minister ma świadomość, ale został złożony projekt dotyczący testowania pracowników domów pomocy społecznej, innych placówek stałego pobytu. Dlaczego nie ma projektu rządowego w sprawie testowania pracowników miejsc, które są najbardziej zagrożone? Niech pani wyciągnie projekt Koalicji Obywatelskiej, proszę z niego skorzystać i proszę się wreszcie wziąć do roboty. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Zwracam się też do nieobecnego na tej sali pana premiera, bowiem pochodzi on z Wrocławia i swego czasu był nawet radnym wojewódzkim, czyli brał odpowiedzialność za losy naszej regionalnej wspólnoty, która jest regionem granicznym sąsiadującym bezpośrednio i z Czechami, i z Niemcami, z Saksonią. Czy wsłuchaliście się państwo w głos protestujących chociażby ostatnio w Zgorzelcu? Oni wznosili następujący okrzyk: zajmijcie się nami, nie wyborami. Nawet gdyby ich było tylko tysiąc, a w skali kraju to jest grubo ponad 100 tys. osób, które nie na skutek fanaberii, ale decyzji rządu nie mogą pracować za granicą w regionach przygranicznych albo są rozdzielone ze swoimi rodzinami, miałyby one prawo oczekiwać, że się nad ich problemem pochylicie. Jeżeli nie potraficie tego zrobić sami, przygotować testów dla tych osób, to pomogą wam (Dzwonek) partnerzy zagraniczni, bo oni również wspierają postulaty Polaków chcących uczciwie pracować, nawet jeśli ta praca wykonywana jest. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Przede wszystkim zdrowie i życie Polaków jest dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego najważniejsze. Wszystkie obostrzenia, które zostały wprowadzone, przede wszystkim służą temu, abyśmy zadbali o zdrowie, o życie Polaków. Przede wszystkim działania, które zostały od samego początku podjęte, pokazują, że są działaniami skutecznymi, które pomagają przez ten trudny czas, w jakim jesteśmy, czas epidemii, przejść jak najbardziej suchą nogą. Te obostrzenia są czasami trudne, natomiast już dziś jesteśmy na etapie pokazywania planowych działań odmrażania gospodarki. I nie są to działania, że my powiemy. Pan premier wyraźnie, pokazując kolejne etapy, nie wskazywał daty, gdyż są one uzależnione od sytuacji epidemicznej, a więc tego, jak te kolejne etapy, w ramach których będziemy to odmrażać, przyczynią się do sytuacji epidemicznej w kraju. Ochrona miejsc pracy zarówno pracowników pracujących w kraju, jak i tych pracujących za granicą jest dla nas wyjątkowa. Przede wszystkim to, co państwo tutaj podnosiliście w swoich wypowiedziach, że tarcze, którym nadajecie numery 1, 2, 3 itd., nie działają, jest nieprawdą.

Możemy śmiało i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że na dzisiaj ochroniliśmy co najmniej 2 mln miejsc pracy.

I takie działania będą przez nas dalej podejmowane. Współpracujemy z samorządami i te samorządy wspieramy. Właśnie współpracujemy, właśnie pomagamy samorządom w tym trudnym czasie.

Przypomnę, że na 824 domy pomocy społecznej na dziś mamy 23 w kwarantannie.

Ale to też było, szanowni państwo.

Pan premier zapowiedział kolejne odsłony, jeżeli chodzi o odmrażanie gospodarki. Powtórzę: nie podajemy konkretnych dat, ale to jest celowe, planowe działanie z tego względu. Ochrona miejsc pracy jest zawarta również w mechanizmach tarczy antykryzysowej.

One przede wszystkim służą Polkom i Polakom oraz polskim rodzinom. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 279) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Romanowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań pozwalających na szybką izolację osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc w sytuacjach, kiedy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Służyć mają temu nie tyle rozwiązania czy zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która obecnie kompleksowo reguluje to zagadnienie, ile zmiany w ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz w ustawie o Policji i w ustawie o Żandarmerii Wojskowej. Jeżeli chodzi o zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, to wprowadzamy tutaj osobny dział w postaci działu dotyczącego rozpoznawania spraw o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Wprowadzamy zatem postępowanie o charakterze odrębnym, które przewiduje szereg uproszczeń zmierzających do przyspieszenia rozpoznawania spraw tego typu. W szczególności są to rozwiązania w postaci nałożenia na sąd obowiązku doręczenia prokuratorowi odpisu wniosku oraz zawiadomienia go o terminach rozprawy, a także rozwiązanie dotyczące możliwości dokonania doręczeń pism przez sąd za pośrednictwem Policji lub Żandarmerii Wojskowej. Określono również terminy do wydania orzeczenia przez sąd oraz terminy do udzielenia zabezpieczenia, tj. odpowiednio 30 i 3 dni, a także wprowadzono natychmiastową wykonalność postanowienia sądowego. Jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o Policji, to projekt wprowadza - i to jest tutaj to istotne rozwiązanie, pierwsze w procesie oddzielania sprawcy przemocy od ofiary przemocy - nowe rozwiązanie, nowe uprawnienie dla Policji w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie i tworzącej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Są uregulowane: sposób zbierania dowodów potwierdzających istnienie przemocy, sposób wnoszenia i rozpoznawania zażaleń, zasady doręczania korespondencji. Przewidziana jest również możliwość przesłuchania przez sąd osób małoletnich. Określony jest czas obowiązywania tych nakazów lub zakazów. Wynosi on 14 dni co do zasady, chyba że zostanie skrócony przez sąd po rozpoznaniu zażalenia, ewentualnie przedłużony w przypadku zastosowania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Jeżeli chodzi o ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, projekt wprowadza rozwiązania analogiczne do tych zastosowanych w przypadku ustawy o Policji co do osób podlegających właściwości Żandarmerii Wojskowej.

Jeżeli chodzi o zmianę w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, w projekcie wprowadza się tryb przyspieszony w przypadku popełnienia wspomnianego wykroczenia. W zakresie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w projekcie wprowadza się zwolnienie osoby dotkniętej przemocą od ponoszenia kosztów sądowych.

Przepis w nowym brzmieniu poszerza dotychczasowe uprawnienia sądu tak, aby były one spójne z uprawnieniami przyznanymi Policji względnie Żandarmerii Wojskowej.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Potrzeba tych zmian jest rezultatem oceny dotychczas obowiązujących przepisów. Polska dołączy do grupy krajów, w których osoby pokrzywdzone przemocą domową uzyskują najlepszą ochronę. Przerywamy w ten sposób pewną spiralę przemocy i milczenia. Bardzo proszę o przyjęcie tych rozwiązań. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Grzegorz Lorek. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 279. Podejmujemy dziś dyskusję nad bardzo ważnym rządowym projektem ustawy, który odpowiada na wyzwania związane z potrzebą wprowadzenia rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc w sytuacji, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Epidemia koronawirusa spowodowała, że w rodzinach, w których wcześniej nie było napięć, mogą one się pojawić. Zostając w domu, każda rodzina musiała się skonfrontować z własnymi mechanizmami radzenia sobie w stanie kryzysu.

Izolacja sprzyja sytuacjom konfliktowym, stresowym, a to może pobudzać agresję osób, które wcześniej nie miały skłonności do stosowania przemocy, i te zachowania eskalować. Przemoc w rodzinie przestała być już postrzegana jako sprawa prywatna, dotycząca jedynie osób stosujących przemoc i dotkniętych przemocą. W sprawie zabrało głos Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało przepisy, o których mówimy, dzięki którym to sprawca przemocy domowej będzie musiał natychmiast opuścić mieszkanie, a osoby pokrzywdzone będą skutecznie chronione. Ustalone zostały także wytyczne dla podmiotów, które w ramach Funduszu Sprawiedliwości wspierają pokrzywdzonych. Organizacje pozarządowe zwracają uwagę na pilną potrzebę zmian legislacyjnych ze względu na rosnącą falę przemocy w związku z izolacją. W tym stanie rzeczy procedowany projekt daje efektywne instrumenty ochrony prawnej osobie doznającej przemocy. Pozwala na wprowadzenie rozwiązań szczególnych dotyczących tej kategorii spraw, które pozwolą sądowi na sprawne przeprowadzanie postępowań. Proponuje się m.in. wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i bezpośredniego otoczenia, co jest bardzo ważne. Umożliwia się sądowi wydanie szczególnego rodzaju postanowienia o zabezpieczeniu oraz doręczeniu orzeczeń sądu i pism sądowych przez policję lub Żandarmerię Wojskową.

Ułatwieniem dla wnioskodawcy związanym z szybkim dostępem do sądu ma być projektowane ustawowe zwolnienie go od kosztów sądowych przewidywanych w nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zupełnie nowym instrumentem mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej przemocą jest dodanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej w zakresie jej właściwości uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i bezpośredniego otoczenia.

Przepisy przewidujące możliwość zastosowania izolacyjnych środków chroniących ofiary przemocy w rodzinie istnieją m.in. w Austrii, której ustawodawstwo stało się wzorcowe dla innych państw. Instrumentami austriackimi służącymi walce z przemocą w rodzinie są m.in. środki zapewniające natychmiastową izolację osoby stanowiącej zagrożenie od ofiary w przypadku stosowania przemocy, nakaz opuszczenia mieszkania, w którym mieszka osoba zagrożona, i jego bezpośredniego otoczenia, nakaz opuszczenia mieszkania i bezpośredniego otoczenia wydany przez sąd. To są regulacje, które już obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Opowiem także, że we Francji wystarczy pójść do apteki, przekazać pewne hasło, które oznacza przemoc domową, i są podejmowane czynności. Projektowane rozwiązania powinny realnie poprawić sytuację osób dotkniętych przemocą. Przyczynią się do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, a także będą pomocne w kształtowaniu prawidłowych relacji między członkami (Dzwonek), przy zachowaniu bezpieczeństwa i godności osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie rekomenduję dalsze procedowanie nad projektem ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Zapraszam, pani poseł. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicja Obywatelska przedstawić stanowisko dotyczące druku nr 279, mowa oczywiście o przemocy domowej. Projekt, który państwo wnieśliście jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest na pewno projektem, który wpisuje się w walkę, jeśli chodzi o przemoc w rodzinie. Wiemy o tym, że tak naprawdę z przemocą domową instytucje państwowe, publiczne rozpoczęły walkę niespełna 20, może trochę przeszło 20 lat temu, ale poprzednie rządy i obecny rząd bardzo różnie podchodziły do problematyki przemocy domowej. Chciałabym przypomnieć, jak wyglądała walka rządów z przemocą domową. Pierwszą fundamentalną ustawą była na pewno ustawa z 2005 r. i tutaj wielką zasługę miała z pewnością pani minister Izabela Jaruga-Nowacka. Kolejną ustawą, która nowelizowała tę ustawę, była ustawa z 2010 r. Wprowadził ją rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To ona zakazywała kar cielesnych w wychowywaniu w rodzinie, to ona wprowadziła zespoły interdyscyplinarne, to ona dawała nowy zakres organizacji, zarządzania „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Naprawdę wiele się zmieniło. Powstawały nowe ośrodki, szły pieniądze do samorządów i to wsparcie dla ofiar przemocy na pewno było lepsze i większe.

Jeszcze gdy trwały prace nad tą ratyfikacją, udało nam się doprowadzić do tego, że gwałt ścigany był z urzędu, a nie na wniosek ofiary.

Polska ratyfikowała konwencję stambulską i na tym tak naprawdę się skończyło. Obecnie urzędujący prezydent na pytanie o konwencję odpowiedział w marcu 2017 r. - najlepiej jej nie stosować. Niestety w 2016 r. słyszeliśmy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwały prace nad wypowiedzeniem tej konwencji, a przecież to, co dzisiaj państwo zaprezentowaliście w tym projekcie, jest właśnie realizacją jednego z postulatów, z postanowień tej konwencji.

To była wasza propozycja skierowana do kobiet, które były ofiarami przemocy w rodzinie. Mało tego, odebraliście pieniądze wielu organizacjom, NGOs, m.in. Centrum Praw Kobiet, które od ponad 20 lat walczyły z przemocą domową, pomagały ofiarom. Tak przez te wszystkie lata wyglądała wasza pomoc ofiarom przemocy domowej. Dzisiaj państwo przynosicie, owszem, dobry projekt i z pewnością go poprzemy. Nie wiem, być może dlatego, że zbliżają się wybory prezydenckie. Chcę państwu powiedzieć, że skorzystamy z tego ukłonu i dzisiaj powiemy wam: sprawdzam, bo boimy się, że ten projekt ustawy ujrzał światło dzienne tuż przed wyborami, ale po wyborach tego projektu może już nie być. Dlatego dzisiaj, pani marszałek, w imieniu klubu Koalicja Obywatelska składam wniosek o niezwłoczne przystąpienie po zakończeniu pierwszego czytania, bez odsyłania projektu do komisji, do dalszego procedowania tego projektu. Zróbmy to natychmiast, tu i teraz, tym bardziej że są szczególne okoliczności i warunki: jest pandemia, są kwarantanny, ofiary są zamknięte ze sprawcami, więc nie ma czasu, nie ma czasu na komisje, nie ma czasu na jakąkolwiek zwłokę. Proszę więc o to, abyśmy jak najszybciej przystąpili do drugiego czytania, bez odsyłania projektu do komisji. Stać nas na to jako opozycję, bo dobre projekty dla ludzi, dla kobiet, dla ofiar (Dzwonek) przemocy, dla słabszych jesteśmy zawsze w stanie poprzeć. Dziękuję bardzo, pani poseł. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica zaprezentuje pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic. Wysoka Izbo! Klub Lewicy zaapelował do pani marszałek Witek o jak najszybsze, niezwłoczne procedowanie nad rządową ustawą umożliwiającą natychmiastową izolację sprawcy przemocy od ofiar. Dziękujemy. O uprawnienia Policji do przerwania katowania i chronienia życia i zdrowia ofiar organizacje kobiece upominają się od lat, a dziś, w dobie pandemii, widać, jak bardzo potrzebujemy tych rozwiązań. Dwa razy dziennie Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Nie informujecie, że Polska jest w ścisłej czołówce Europy w liczbie samobójstw dzieci poniewieranych także przez ich najbliższych. Nie informujecie, bo to wstyd, że państwo w centrum Europy nie jest w stanie zagwarantować ludziom elementarnego bezpieczeństwa, oferując jedynie slogany o świętości polskiej rodziny i cierpieniu, które ponoć uszlachetnia. Zostań w domu - mówicie. W domu, który bywa miejscem kaźni, gwałtów, bicia, poniewierania. 30% - o tyle wzrosła przemoc domowa w krajach, które wprowadziły samoizolację, bo kryzys rodzi frustrację, a frustracja musi wybuchnąć. O ile więcej jest cierpienia, skoro rządowe statystyki mówią o prawie 100 tys. ofiar przemocy domowej rocznie, a badania naukowe mówią, że to 10. część prawdziwej skali zjawiska? Te wszystkie domowe tragedie i śmierci wydarzyły się nie z powodu obojętności sąsiadów, ale obojętności kolejnych rządów na problem przemocy w rodzinie. Kiedy pan, panie ministrze Ziobro, obejmował w 2015 r. stanowisko ministra, przejmował pan odpowiedzialność, dosłownie, za prawo i sprawiedliwość - za prawa wszystkich pokrzywdzonych przez przestępstwo i za sprawiedliwość dla sprawców i ofiar. A pierwsze, co pan zrobił, to był skok na fundusz zwany przez was, chyba sarkastycznie, Funduszem Sprawiedliwości. Zabraliście dotacje organizacjom pomagającym kobietom i dzieciom o największym dorobku i osiągnięciach, bo nie podobały się wam ich równościowe poglądy. Na niektóre nasłaliście policję i unurzaliście je w błocie aluzji i obrzydliwych sugestii. I po co to było, skoro koniec końców przyznaliście im wszystkim, nam wszystkim rację, że sprawcę trzeba natychmiast izolować i że prawo do życia i bezpieczeństwa jest ważniejsze niż domowy komfort agresorów? Kilka dni temu miliony, które mogłyby być przeznaczone na pomoc pokrzywdzonym, poszły z ministerialnej kasy na fundację księdza egzorcysty, księdza, który, cytuję, walczy z demonami wegetarianizmu, a do egzorcyzmów używa salcesonu. Będziecie egzorcyzmować katowanych i poniewieranych? Co to ma być? Ministerstwo Sprawiedliwości czy ministerstwo śmiesznych kroków? W południowej części Lubuskiego w pierwszym roku waszych rządów udzielono pomocy 4-, 5-krotnie mniejszej liczbie osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa niż rok wcześniej. To był skutek tego skoku. Ówczesna ministra pracy, rodziny i polityki społecznej opowiadała, że 500+ rozwiązuje problem przemocy domowej, bo bite kobiety mogą się wyprowadzić. Faktycznie, doskonały pomysł, zwłaszcza w dzisiejszych realiach. A „Niebieskiej karty” nadal nie można wypełnić zdalnie. Dlaczego? A co zrobiliście dla bitych dzieci, bitych właśnie w tej chwili, które nie chodzą do szkoły i nie mają komu powiedzieć, że ojciec czy matka je katują? Koronawirus obnażył wszystkie zaniechania waszego rządu. Zajął się pan, panie ministrze, przejmowaniem władzy nad prokuraturą i sądami, żeby po 5 latach przyznać, że ani ministerialne fundusze, ani sądy czy prokuratura nie są skuteczne w ratowaniu kobiet i dzieci, że musi to robić Policja, która panu nie podlega. Od 20 lat codziennie patrzę w moim stowarzyszeniu BABA na twarze bitych ludzi. Patrzyłam w oczy ojca, którego córka podcięła sobie żyły, bo gwałcił ją dziadek. Patrzyłam w oczy dzieciom, których ojciec zakatował matkę. Chcę tym ludziom spojrzeć w oczy i powiedzieć, że Sejm uznał ich życie i bezpieczeństwo za ważniejsze niż liczenie szabel Gowina. Procedujmy, czas ucieka, tik-tak, tik-tak. Niejedną ustawę przyjęto tutaj ekspresowo, w ciągu kilku godzin. Dziś i jutro zginą trzy kobiety. Dziś, jutro, najdalej w piątek rano zabije się katowane dziecko. Niech prezydent ekspresowo to podpisze. Jeszcze zdąży zrobić coś dobrego, nim straci władzę. Tylko niech upływającego czasu nie pomyli z TikTok. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 głos zabierze pani poseł Agnieszka Ścigaj, zdalnie. Wiem, że już mamy połączenie, tak? Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 dotyczące projektowanej ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 279. Ustawa dotyka bardzo poważnego zjawiska, takiego zjawiska, które rzeczywiście w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj, niestety się nasila. Wszystkie dane statystyczne wskazują na to, że nie tylko nasila się i wzrasta przemoc w rodzinach, które były już zdiagnozowane i rozpoznane jako te, które tę przemoc stosowały, ale również pojawiają się nowe rodziny, nowe sytuacje. Sytuacja konfliktowa, sytuacja utraty poczucia bezpieczeństwa na każdym poziomie, każdego obywatela niestety wiąże się z tym, że wyzwala złe emocje. Niestety tak się dzieje i w tych dniach mamy te dane takie, jakie mamy. Ustawa jest bardzo dobra, to ustawa, którą proponowały środowiska organizacji pozarządowych zajmujących się od lat przemocą. Ustawa, która od wielu, wielu lat z powodzeniem istnieje i funkcjonuje w innych państwach i rzeczywiście skutecznie chroni ofiary. Sprawca się panoszył, a ona latami dochodziła swoich praw, bardzo często przed sądem, samotna. To jest wreszcie krok w dobrym kierunku. My jesteśmy gotowi poprzeć tę ustawę, ale jednocześnie apelujemy - ponieważ ta ustawa jest tylko rozwiązaniem prawnym absolutnie koniecznym i jesteśmy, tak jak pozostałe kluby, za tym, żeby nad nią procedować natychmiast - że w tarczy, nad którą w tej chwili procedujemy, ważne jest, żeby dojść do sytuacji, że nie tylko sama izolacja i szybka reakcja jest potrzebna, ale przede wszystkim wsparcie psychologiczne, wsparcie psychiatryczne.

Trzeba tym rodzinom pomagać, trzeba pomóc dzieciom, ktoś te rodziny musi odwiedzać.

I tak jak wcześniej mówiliśmy, wszystkie dobre projekty, które państwo składacie, będziemy popierać, a wszystkie złe będziemy krytykować. I ważne, żeby na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych również podjąć dyskusję, żeby do tarczy nr 3, którą państwo proponujecie, wprowadzić dodatki i odpowiednie środki dla pracowników pomocy społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Żeby nie zapomnieć, w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja wnoszę o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego naprawdę głęboko złego projektu. Nie leczmy dżumy cholerą, szanowni państwo.

Ta infekcja, ta franca, szanowni państwo, szerzy się w ten sposób: najpierw generuje się katastrofę społeczno-gospodarczą, a potem leczy się objawowo na bardzo różne sposoby. Najpierw, żeby nie sięgać głębiej, aż do bismarckowskich Prus i innych pożałowania godnych wzorców, przykład z ostatnich czasów, z ostatnich chwil. Chodzi o tu przez państwa wzmiankowane pierwotne przyczyny tego doraźnego zła. Zamknijcie ludzi w mieszkaniach, nie pozwólcie im wychodzić na wiosenne słoneczko, żeby nabywali naturalnej odporności i dotleniali się, dzięki czemu człowiek od razu lepiej funkcjonuje. Zamknijcie ich tam i wygenerujecie problemy społeczne, jasna sprawa. Wzorce zagraniczne. Austria. No nie, dziękuję. To są wzorce które.

Australia, na tę samą literę. Jeśli już chcecie majstrować przy rodzinie, szanowni państwo, to w Australii jest taki oblig prawny, że zwołuje się de facto radę familijną. Mówię to, pochylając się z troską nad wszystkimi przypadkami, które wypada potępić, i Konfederacja potępia je. My, państwowcy, ludzie stojący twardo na gruncie tradycyjnie pojmowanych zasad cywilizacyjnych prawa, rzecz jasna, nie możemy inaczej patrzeć na złoczyńców niż jak na delikwentów, których trzeba stawiać przed sądami, niezależnie od płci notabene, niezależnie od tego, czy to są damscy bokserzy, czy to są krewkie niewiasty tłukące mężczyzn, którzy też gdzieś tam, po domach, cierpią w cichości. Ale powiadam: sprowadzać wszystkim od razu na kark żandarma, policjanta, to jest leczenie dżumy cholerą. Konwencja stambulska - ależ tak, właśnie ją należy jak najszybciej wypowiedzieć. Ależ tak! Ona bowiem stygmatyzuje rodzinę jako taką, wskazuje oskarżycielskim paluchem, rządowym niestety, rodzinę jako matecznik zła, generator tragedii, a nie ciągłości tradycji. Potępiajmy, ścigajmy i nie wahajmy się karać przykładnie przestępców, ale nie twórzmy mechanizmu, który będzie kolejną.

Można z tego zacząć korzystać jako z udatnych pretekstów do tego, żeby pogłębiać tę ingerencję. Wniosłem zatem o odrzucenie tego niedobrego projektu i wnoszę o to, także i przy tej okazji, żebyście państwo wsłuchali się we własne głosy, żebyście cofnęli i przewinęli taśmę, żebyście usłyszeli, jak mówicie o fatalnych przyczynach pozostawania ludzi w zamknięciu, kiszenia się po domach. Nie generujcie katastrofy gospodarczej, za którą musi iść katastrofa socjalna, upadek - tak jest - moralności. Na to tu za mało jest państwa, żeby słychać było dostatecznie głośno buczenie, ale słyszę, że buczycie wewnętrznie. Tak, trzeba wracać do korzeni, do tradycji, a nie leczyć objawowo.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Informuję panie i panów posłów, iż Prezydium Sejmu na podstawie art. 39 ust. 1 regulaminu Sejmu ustaliło w tym punkcie limit 30 pytań dla klubów według następującego parytetu: Prawo i Sprawiedliwość - 15, Koalicja Obywatelska - 9, Lewica - 3, PSL-Kukiz15–2, a także jedno pytanie dla koła. Zamykam listę. Zapraszam.

Wysoka Izbo! Są mordowane przez swoich partnerów, umierają w wyniku pobicia albo popełniają samobójstwo. O ten projekt ustawy, nad którym dzisiaj procedujemy, od lat zabiegają organizacje pozarządowe, rzecznik praw obywatelskich.

Fundacja BABA, Centrum Praw Kobiet, Niebieska Linia, Amnesty International i wiele, wiele innych organizacji, osób prosiło, błagało, apelowało, mówiło o tym, że konieczna jest izolacja oprawcy od ofiary, że to nie na ofierze musi spoczywać obowiązek zadbania o swoje bezpieczeństwo w obliczu tak strasznej tragedii, jaką jest przemoc domowa. To jest dobra zmiana, nad którą trzeba procedować natychmiast, bo niestety dotychczasowa polityka Prawa i Sprawiedliwości była wyznaczona przez Beatę Szydło, która chwaliła jedyną gminę w Polsce (Dzwonek), która nie wdrożyła ustawy antyprzemocowej. Zróbmy to jak najszybciej. Bardzo proszę. Szanowny Panie Ministrze! Od 20 lat kobiety i środowiska kobiece domagają się kompleksowych regulacji dotyczących ochrony kobiet przed przemocą i przeciwdziałających tej straszliwej patologii życia społecznego. Sprawna, szybka i skuteczna izolacja sprawcy przemocy od ofiary to standard, o który organizacje kobiece broniące praw kobiet zabiegają od lat. Dzięki niej wiele kobiet mogłoby uratować swoje życie przed zwyrodnialcami i nie musiałoby uciekać z dziećmi z domu, by tułać się po przytułkach. Dlatego też chciałabym zapytać pana ministra, czy rząd rzeczywiście ma zamiar jak najszybciej procedować nad tą ustawą, która wprowadza silne instrumenty prawnej ochrony kobiet i ich rodzin, o co wnioskuje Lewica. Czy rzeczywiście chcecie jak najszybciej pomóc kobietom?

Bardzo proszę.

Państwo prześledźcie ten łańcuch przyczynowo-skutkowy, nie leczcie objawowo. Najpierw fundujecie Polakom niewydolne sądy, a potem rozglądacie się za procedurą, która przyspieszy ich działanie. Najpierw wprowadzacie przykrą dla samych funkcjonariuszy uznaniowość w ich działaniu - areną takich spektakli i śmiesznych, i strasznych jest Rzeczpospolita w ostatnich tygodniach - a potem musicie to wszystko uściślać, porządkować pod pretekstem, nie daj Boże, walki z jakimś wrażym wirusem, mniemaną pandemią. To jest właśnie świat żoliborskich socjalistów, gdzie rozwiązuje się bohatersko problemy, które nie byłyby znane w normalnym świecie, czyli w takim świecie, który nie odrywa narodu polskiego od pnia cywilizacyjnego (Dzwonek), od autentycznych źródeł praworządności, sprawiedliwości. Pytanie: Kiedy wypowiecie konwencję stambulską i czy sprawa jest na warsztacie? Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Koleżanki i Koledzy Posłowie! Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie musi być skuteczna, a nie tylko zadeklarowana na papierze. Jednym z podstawowych warunków jej skuteczności jest m.in. szybkie izolowanie sprawcy od ofiar. Dlatego z zadowoleniem, panie ministrze, ten projekt witam i wiem, że te 90 tys., według oficjalnych danych, ofiar przemocy w rodzinie czeka na ten projekt. Jednak rzeczywiście, tak jak tutaj mówiły już moje przedmówczynie, nie byłoby tego projektu, gdyby nie lata walki organizacji pozarządowych. Pierwsza z nich to Centrum Praw Kobiet, które ponad 20 lat temu rozpoczęło właśnie walkę z przemocą w rodzinie, często było wyśmiewane. Ale tak jak powiedziałam, prawo to jedno, natomiast to prawo musi być skuteczne.

Szkolenia policjantów i Żandarmerii Wojskowej.

Mam nadzieję, że z Funduszu Sprawiedliwości doczekają się wsparcia te organizacje pozarządowe, które od lat walczą z przemocą, z tym strasznym zjawiskiem, a nie tylko takie organizacje jak wspomniana już tutaj fundacja założona przez byłego egzorcystę. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Projekt ustawy, nad którym procedujemy, może uratować życie i ochronić zdrowie wielu kobiet i dzieci w Polsce. Dlatego niezwłocznie powinniśmy przystąpić do kolejnego czytania, przyspieszając uchwalenie i wejście w życie tych ważnych przepisów. Zbyt długo, pomimo apelu różnych środowisk, musieliśmy czekać na przepisy umożliwiające skuteczną izolację sprawców przemocy. Ustawa to jedno, a rzeczywistość jest brutalna. Przy moim biurze poselskim w Kielcach działa świętokrzyskie Centrum Praw Kobiet. Pracownicy codziennie odbierają telefony od maltretowanych ofiar przemocy domowej. Dochodzi do dramatycznych przypadków, że policja, przyjeżdżając z interwencją, wprost informuje, jak dużo ma pracy w związku z pandemią, a kolejne wezwanie może zostać ukarane mandatem. Nagminnie łamany jest sądowy zakaz zbliżania się. Przez bezczynność rządu od lat Polska jest ogarnięta inną epidemią: bitych i prześladowanych psychicznie kobiet i dzieci. Dlatego najwyższy czas na zmiany. Czas na zdrową Polskę (Dzwonek) i nową nadzieję dla kobiet i maltretowanych osób. Pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od dawna apeluję o nadzwyczajne środki ochrony ofiar przemocy. Teraz, w czasie powszechnej izolacji, one są szczególnie istotne. Wiele zapisów w tym projekcie należy uznać za słuszne, jednak ważniejsze jest pytanie, czy za tymi przepisami pójdą konkretne działania pomocowe ministerstwa, czy organizacje wspierające ofiary przemocy dostaną dodatkowe środki i czy będą mogły skutecznie pomagać. Widać skokowy wzrost liczby próśb o interwencję, np. na „Niebieską linię” Biorąc pod uwagę tylko kwiecień, jest 70% więcej zgłoszeń mailowych. Te zgłoszenia są bardziej emocjonalne, one są wręcz dramatyczne.

Pamiętamy, jak państwo chcieli legalizować przemoc, mówiąc, że jedno pobicie to nie jest przemoc. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przemoc domowa w Polsce ma charakter systemowy i głęboko zakorzeniony w naszej kulturze i tradycji. Powiedzenie: jak chłop baby nie bije, to jej wątroba gnije, nie wzięło się znikąd. Niestety zbyt często dokłada się do tego polski Kościół katolicki, mówiąc maltretowanym kobietom z ambon albo w konfesjonałach: rodzina jest święta, musisz nieść swój krzyż. Kilka lat temu minister sprawiedliwości Jarosław Gowin nie chciał podpisania konwencji antyprzemocowej, bo niby zagraża polskiej tradycyjnej rodzinie, gdyż zobowiązuje państwa do wykorzenienia uprzedzeń i złych zwyczajów i tradycji. Dobrze, że rząd chce pomóc ofiarom przemocy i izolować sprawców. Ale jak rząd chce edukować przeciw przemocy? Jak chce zwalczać przyczyny przemocy?

Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ustawa jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że jak najszybciej wejdzie w życie. Pierwsze. Wiele słyszy się w opinii publicznej na temat przepełnionych noclegowni czy schronisk dla bezdomnych. Projekt procedowanej ustawy zakłada, iż do takich miejsc nakazem Policji zostanie przekazany sprawca przemocy domowej. Gdzie zostanie ulokowany oprawca w momencie, kiedy wszystkie miejsca noclegowe będą zajęte? Czy macie państwo jakąś alternatywę? Kto zapewni transport takiej osoby np. do sąsiedniej miejscowości, jeśli tam znajdzie się wolne miejsce? W jaki sposób Policja będzie weryfikowała potencjalnych oprawców? Czy jedno zgłoszenie wystarczy, aby sprawca przemocy domowej otrzymał nakaz opuszczenia miejsca zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym? Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! W końcu bite kobiety, maltretowane dzieci doczekały się projektu ustawy, który daje im poczucie bezpieczeństwa we własnym domu, który daje Policji możliwość odizolowania sprawcy przemocy natychmiast, bez sądów, bez procedur, tak aby mogły spać spokojnie. Zastanawia tylko, dlaczego tak późno i dlaczego teraz. Bo jest problem, szanowni państwo. Mój niepokój budzi fakt kwalifikacji czynu. Czyn ten w momencie złamania przez sprawcę zakazu, nakazu wydanego przez Policję jest kwalifikowany jako wykroczenie. Dlaczego? Są zbyt niskie kary dla oprawców i sprawców przemocy domowej. Powinny być restrykcje takie, które dają poczucie bezpieczeństwa rodzinie, matkom i dzieciom. Pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mamy trudny czas, ważny projekt i bardzo delikatny obszar dotyczący ochrony ofiar przemocy. Moje pytanie wynika z troski o małoletnie dzieci wychowywane przez sprawców przemocy domowej. Projekt ustawy zakłada natychmiastowe opuszczenie lokalu mieszkalnego przez oprawcę. Jak będzie wyglądała procedura opuszczenia lokalu, w przypadku gdy oprawcą jest osoba samotnie wychowująca dzieci? To powinno nas szczególnie interesować, bo dzieci wyciągnięte z domowego piekła mogą zostać wepchnięte w inną traumę. Kto zaopiekuje się tymi dziećmi? Jak będzie wyglądał proces przejęcia opieki nad małoletnimi? Czy rząd planuje przeszkolić funkcjonariuszy Policji czy Żandarmerii Wojskowej w zakresie postępowania z pokrzywdzonymi małymi dziećmi - ofiarami przemocy? Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przemoc w rodzinie to nie jest sytuacja wyjątkowa, lecz niestety brutalna codzienność. Tylko z oficjalnych zgłoszeń wynika, że rocznie ofiarami przemocy jest blisko 90 tys. osób, a 3/4 ofiar to kobiety. W tej sytuacji nie można zapomnieć, że od lat konsekwentnie robicie wszystko, żeby pozbawić te ofiary wsparcia. Przypomnę tylko: to wasz upartyjniony prezydent mówił, żeby konwencji antyprzemocowej nie stosować, to wasz rząd konsekwentnie odmawia dofinansowania organizacjom, które walczą z przemocą, i nie przyznał dotacji, np. na „Niebieską linię” Dlatego chciałbym zapytać: Kiedy rząd zmieni swoje podejście, tak żeby osoby doświadczające przemocy mogły otrzymać rzeczywiste wsparcie i czuły się w Polsce bezpiecznie? W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim organizacjom feministycznym, dziecięcym, LGBT+ i rzecznikowi praw obywatelskich, wszystkim, którzy dzień w dzień ciężko pracują (Dzwonek), żeby pomóc ofiarom przemocy. To dzięki nim ten projekt dzisiaj jest procedowany. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszę się, że debatujemy dzisiaj nad projektem ustawy w tak ważnej kwestii, jak ochrona osób dotkniętych przemocą domową, poprzez ich szybką i skuteczną izolację od osób stosujących przemoc. Cieszy mnie to, że tym projektem realizujemy art. 53 konwencji stambulskiej, konwencji, którą wnioskodawcy wielokrotnie zapowiadali wypowiedzieć. Artykuł ten zobowiązał nas do przyjęcia koniecznych środków do zapewnienia ofiarom przemocy domowej możliwości wystąpienia o odpowiednie nakazy i zakazy ochronne, co też ten projekt ustawy czyni. Cieszy mnie to, że nareszcie korzystacie z dorobku organizacji kobiecych, którym jeszcze tak niedawno obcinaliście publiczne finansowanie. O ile ten projekt jest krokiem w dobrą stronę, to mam jednak kilka pytań dotyczących obecnych działań. W tej chwili przemoc w domach nasila się ze względu na bardzo trudną sytuację, izolację i zamknięcie. W jaki sposób Policja (Dzwonek) i władze publiczne zapewniają bezpieczeństwo osobom narażonym na przemoc?

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Panie Pośle! Przedstawione założenia zmiany Kodeksu karnego i działania to właściwy krok w bardzo dobrym kierunku. Przyjmujemy to jako coś, co ma zapowiedzieć kompleksową opiekę nad ofiarami przemocy domowej. Należy natychmiast separować sprawcę przemocy od ofiar, często dzieci i kobiet.

Po interwencji osobom, głównie kobietom, dzieciom, często także starszym rodzicom, trzeba pomóc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. To są często bardzo traumatyczne wybory, związane z kontynuacją pracy i edukacji.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Marcin Romanowski. Zapraszam, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o zagadnienia, które zostały poruszone, to warto zwrócić uwagę na historię tego projektu.

To niewątpliwie bardzo trudne i kompleksowe zagadnienie wymagało szerokich badań i analiz. Chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście, jak tutaj było podnoszone, postulat dotyczący wprowadzenia tego typu rozwiązań pojawiał się już od wielu lat, od kilkunastu lat. Jak tylko przyszliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości, rozpoczęliśmy nad nim pracę. Rodzi się pytanie: Dlaczego ten postulat nie został zrealizowany wcześniej, kiedy rządziły Platforma Obywatelska i PSL przez 8 lat, wtedy on był również podnoszony? Wydaje mi się, że odpowiedź jest taka, że my nie zajmujemy się ideologią, tylko rozwiązywaniem realnych problemów osób pokrzywdzonych przestępstwem i realnym ściganiem sprawców tych przestępstw, domniemanych sprawców - nie ideologią. Myślę, że to jest odpowiedź na wiele uwag i komentarzy. Chciałbym też zwrócić uwagę, że w naszej ocenie jest to rozwiązanie niezbędne, aby chronić rodzinę, aby rodzina, która jest ważną podstawową komórką społeczną, rzeczywiście pełniła swoją doniosłą rolę, której żadna instytucja nie jest w stanie zastąpić. Ale po to, żeby tak było, konieczne są tego typu rozwiązania. W naszej ocenie przemoc nie ma barw ideologicznych czy politycznych, nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, jest po prostu przemocą. Należy ją zwalczać. To jest w naszej ocenie rozwiązanie, które w tym momencie stanowi dopełnienie systemu, bez którego ten system, który funkcjonuje od lat, jest niewydolny.

Przypomnę, że w zeszłym roku zostały wprowadzone rozwiązania dotyczące generalnie postępowania cywilnego, również rozwiązania o charakterze specjalistycznym, takie jak właśnie sądy własności intelektualnej. Ten projekt dotyczy również usprawnienia postępowania w ramach procedury cywilnej poprzez wprowadzenie postępowania odrębnego. Doświadczenie pokazało, że było to nieskuteczne. My to przeanalizowaliśmy i zaproponowaliśmy zmianę, która w naszej ocenie będzie realną i skuteczną zmianą.

W naszej ocenie jest to możliwe.

Ono znalazło się w ustawie o Policji również dzięki bardzo dobrej współpracy z ministerstwem spraw wewnętrznych, za którą chciałbym też przy tej okazji podziękować. Myślę, że formularze policyjne, które na tej podstawie będą realizowane, mają teraz bardzo dobrą podstawę ustawową i podstawę, która wynika z wieloletniego doświadczenia. Jeżeli chodzi przy okazji o szkolenia, to tak, już byliśmy na etapie przygotowywania tego projektu, na etapie uzgodnień międzyresortowych w kontakcie z ministerstwem spraw wewnętrznych i Ministerstwem Obrony Narodowej. Przygotowujemy, już jesteśmy w trakcie przygotowywania kompleksowych szkoleń, jeżeli chodzi właśnie o Policję (Dzwonek) i Żandarmerię Wojskową. Jeżeli chodzi o lekarzy sądowych, to pozwolę sobie odpowiedzieć pisemnie, ze względu na czas. Dodam, że w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości po raz pierwszy stworzyliśmy kompleksową sieć pomocy osobom pokrzywdzonym. Mamy tam rozwiązania dotyczące kompleksowej pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, również materialnej, która to sieć będzie również zastosowana do wsparcia i realizacji tej ustawy. Przewidzieliśmy rozwiązania, które nie tylko wskazują na obowiązek Policji polegający na poinformowaniu o możliwości skorzystania z pomocy, ale przewidujemy nawet możliwość czy takie rozwiązanie, które polega na tym, że dane osoby pokrzywdzonej przez przemoc w momencie zastosowania nakazu policyjnego będą przekazane wprost do ośrodków pomocy pokrzywdzonym, chyba że ta osoba oczywiście wyrazi sprzeciw. Tutaj nie wprowadzamy zmian w zakresie procedury karnej, tylko procedury cywilnej, więc chodzi o naruszenie pewnego nakazu czy orzeczenia sądu. Nie zmieniamy w ogóle rozwiązań o charakterze prawnokarnym. Jeżeli chodzi o kwestie pozostawienia, mówiąc krótko, dzieci bez opieki, to tutaj oczywiście będą miały zastosowanie normalne regulacje dotyczące kwestii opieki nad dziećmi. Jeżeli chodzi o kwestie lekarskie, to odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz wnioski o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk nr 300) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju pana Krzysztofa Mazura o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jak państwo wiecie, od początku zmagania się z pandemią nasz rząd uruchamia szereg instrumentów, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom.

Oprócz tego uruchomiliśmy również poza tą pierwszą i drugą tarczą tarczę finansową. Tu Polski Fundusz Rozwoju uruchomił mechanizmy, które dzisiaj od godz. 18, czyli za 15 minut, będą uruchomione. W tych wszystkich działaniach chodziło o szybkość, chodziło o to, żeby jak najszybciej pomoc trafiła do potrzebujących.

To jest działanie, które nie ma charakteru szybkiej interwencji, szybkiej pomocy, tylko jest nastawione na strukturalną pomoc tym firmom, które będą miały na tyle poważną sytuację, że będą potrzebowały głębokiej restrukturyzacji.

Co istotne, proponowana ustawa jest zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. To oznacza, że skoro jest inna podstawa europejska dla tej pomocy, to ta pomoc nie będzie sumowała się z tą, która jest udzielana w tych instrumentach, które już zostały uruchomione. Czyli jeżeli jakaś firma otrzyma w ramach tarczy antykryzysowej czy tarczy finansowej pomoc, to ta pomoc nie będzie się sumowała.

Jak powiedziałem: to jest długoterminowa pomoc, nawet do 10 lat, i może wynosić nawet do 10 mln euro na jedną firmę. Jakie instrumenty proponujemy? Proponujemy tak naprawdę trzy typy instrumentów, trzy typy pomocy. Po pierwsze, krótkookresowe pożyczki. To są pożyczki do 6 miesięcy. Jeśli to okaże się niewystarczające, to mogą one być przesunięte na kolejne 18 miesięcy. To są krótkookresowe pożyczki, które mają na celu przede wszystkim utrzymanie płynności. Chodzi o zastanowienie się, na ile firma wyjdzie z kłopotów, a na ile będzie musiała przejść restrukturyzację. Jeśli okazałoby się, że ona potrzebuje dalszej restrukturyzacji, to mamy krok drugi, i to jest tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. To jest kolejne 18 miesięcy, kiedy firma w kłopotach może otrzymać od nas pomoc i korzysta z tej pomocy, przeprowadzając plan restrukturyzacji na własną rękę. To jest to narzędzie, które jest nazywane pomocą na restrukturyzację.

Dzięki temu ta firma może wyjść z kłopotów. Co w ramach tego planu restrukturyzacyjnego? Oprócz pożyczki dostępne są również wejścia kapitałowe oraz ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. To ma na celu przygotować rzeczywiście taką pomoc tym firmom, żeby nawet przy głębokiej restrukturyzacji były one w stanie przetrwać, zmieniając swój profil działania, dalej funkcjonować. Tak że, tak jak powiedziałem, jest to długofalowe działanie po tym krótkofalowym działaniu związanym z tarczą.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tej ustawy, gdyż wydaje nam się, że po tych działaniach doraźnych, których celem była jak najszybsza pomoc przedsiębiorstwom, potrzebujemy właśnie takiej ustawy, która będzie długofalowo, przez 10 lat prowadziła firmy poprzez restrukturyzację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zabierze pan poseł Przemysław Czarnek, zdalnie. Wiem, że już jest połączenie. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Mam zaszczyt przedstawić stanowisku klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

To prawda, że instrumenty wsparcia z tarczy antykryzysowej mają charakter krótkoterminowy i z założenia mają być i są natychmiastowo dostępne tu i teraz, wbrew tym wszystkim głosom, które dzisiaj w trakcie dyskusji nad innymi punktami słyszeliśmy. Mogę podać przykłady, o które prosiła pani marszałek Kidawa-Błońska, sugerując, że nikt wsparcia od rządu nie dostaje, i chciałaby przykładów z imienia i nazwiska. Mogę je podać, jestem w kontakcie bezpośrednim z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy panem Andrzejem Pruszkowskim w Lublinie.

To jest tylko przykład tego działania tu i teraz.

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców jest przewidziany jako działanie uzupełniające dla tarczy antykryzysowej i następujące po zastosowaniu instrumentów tarczy.

Projekt ustawy tworzy instrumenty wsparcia, które mają zapewnić przedsiębiorcom płynność finansową na czas przygotowania działań naprawczych i umożliwić sfinansowanie tych działań w ramach przygotowanego planu restrukturyzacyjnego. Formy, które zostały zaproponowane, a zatem nakierowane na ratowanie, a także tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, powinny być w naszym przekonaniu jak najszybciej dostępne dla właścicieli firm jako komplementarne, uzupełniające tarczę antykryzysową wsparcie długoterminowe. Dlatego też klub Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za dalszymi, sprawnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Waldemar Sługocki.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawić stanowisko klubu wobec projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Bardzo mnie cieszy to, iż mój przedmówca tak pozytywnie odniósł się do tego projektu ustawy, gdyż - przypomnę - wpisuje się on w „Politykę nowej szansy”, politykę, która została uchwalona przez parlament 22 lipca 2014 r. i jest autorstwa naturalnie koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe - Platforma Obywatelska. Owszem, trzeba dodać, że jest to instrument długoterminowy, ale jest to instrument, proszę państwa, który moim zdaniem będzie instrumentem, który nie będzie w ogóle terminowy, ponieważ gros polskich podmiotów gospodarczych nie będzie mogło z niego skorzystać pomimo bardzo ważnych i istotnych celów, jakie zostały w tym projekcie ustawy zapisane. Po pierwsze, trzeba zacząć od tego, proszę państwa, że czas, w którym procedujemy nad tą ustawą, jest absolutnie niezadowalający, i to niezadowalający ze strony polityków opozycji czy też polityków opcji rządzącej, ale przede wszystkim jest niezadowalający, ponieważ czekają na to wsparcie polscy przedsiębiorcy, którzy bardzo ciężko znoszą zamrożenie polskiej gospodarki. Przypomnę, że podstawa prawna do uruchomienia pomocy publicznej sięga roku 2015.

W Polsce pierwszy pacjent zero pojawił się w dniu 4 marca w Zielonej Górze. Projekt ustawy, który nie tylko nie wpisuje się, jeżeli chodzi o przedział czasu, ale także, w mojej ocenie, jest niezwykle trudny z punktu widzenia barier administracyjnych. Jeżeli państwo dokładnie przeanalizujecie formę oraz ilość załączników, jakie są zobowiązane przygotować poszczególne podmioty gospodarcze, to zauważycie, że skala dokumentów, przygotowanych materiałów jest tak wielka, że gros podmiotów gospodarczych będzie miało z nimi niezwykle duże problemy.

Otóż minister właściwy do spraw gospodarki czy też podmiot przez niego wskazany, polska agencja rozwoju, ma 30 dni na zweryfikowanie dokumentów, w uzasadnionych przypadkach - do 45, po czym beneficjent, biorca, aplikant tychże środków finansowych ma 7 dni na odniesienie się ewentualnie do sugestii tychże instytucji, po czym, proszę państwa, ewentualnie następne 30 dni na sformułowanie odwołania wtedy, kiedy ten projekt zostanie oceniony negatywnie. Natomiast instytucja, która przydziela i decyduje, podejmuje de facto decyzję o przyznaniu tych środków, ma 60 dni na udzielenie odpowiedzi.

Niepokoi to, szanowni państwo, że pan premier Mateusz Morawiecki z wielką niechęcią i w sposób skrajnie negatywny mówi o Unii Europejskiej.

W imieniu klubu Lewica głos zabierze pan poseł Adrian Zandberg. Bardzo proszę. Nie ma pana posła.

Wysoka Izbo! Czasy przyszły wyjątkowe i wróciły w tej Izbie słowa, których dawno tu nie było: zwolnienia grupowe, masowe bezrobocie, cięcia, wreszcie restrukturyzacja. W takim czasie wyjątkowa staje się odpowiedzialność państwa. Opowieść o tym, że rynek dobrze sobie radzi bez pomocy państwa, brzmiała dobrze podczas prosperity, ale jak zawsze okazała się niewiele warta w chwili próby. Pomoc dla przedsiębiorstw, które są dziś zagrożone upadłością, jest konieczna. Ale muszę powiedzieć, że uśmiechałem się pod nosem, czytając tę ustawę, bo miałem poczucie, że to jest produkt z przeszłości, wręcz zamierzchłej przeszłości, bo wszystko teraz, w czasie kryzysu, dezaktualizuje się naprawdę szybko. I nic dziwnego, bo oczywiście powinniście byli państwo to narzędzie uruchomić już dawno temu.

Niestety jest jeden problem: środki, które zapisaliście w tych przepisach, mogą wywołać co najwyżej wzruszenie ramion, bo 120 mln zł to są pieniądze zupełnie niewspółmierne do skali problemów, z którymi będziemy się borykać, wychodząc z tego kryzysu. On jest zbyt skromny, żeby realnie kryzys zamortyzować. Mówimy tu o wydawaniu publicznych środków, a w związku z tym trzeba bardzo uczciwie porozmawiać o celach i o warunkach tej pomocy. I tego niestety w tej ustawie mocno brakuje. Nie wolno powtórzyć błędów z przeszłości, kiedy uspołeczniono straty, a zyski trafiły do nielicznych kieszeni najbogatszych. Dlatego Lewica zgłosi do tego projektu konkretne poprawki. Tam gdzie płynie pomoc, powinien obowiązywać kategoryczny zakaz wypłaty premii i bonusów, dodatkowych bonusów dla kadry zarządzającej. Niestety po wprowadzeniu waszej antypracowniczej tarczy już związkowcy donoszą, że kolejne zarządy obcinają pracownikom płace, ale swoim członkom wynagrodzenia podnoszą. Ale to też dowodzi, że pomoc musi być realnie kontrolowana, inaczej zamiast na ratowanie firm, zamiast na ratowanie miejsc pracy w rzeczywistości trafi do prywatnych kieszeni nielicznych. Jeżeli ktoś sięga po publiczne środki, to znak, że czas obscenicznych wynagrodzeń dla zarządów tej firmy się skończył, i najwyższy czas, żeby to jasno powiedzieć. Te pieniądze mają służyć utrzymaniu działalności, a nie utrzymaniu luksusowego życia panów prezesów. I oczekujemy wprowadzenia takich zmian, które przed tym zabezpieczą. Wreszcie sprawa kluczowa - warunki zatrudnienia, obowiązek zatrudniania na uczciwych warunkach. Firmy, które przetrwają przy pomocy państwa, dzięki pomocy państwa, nie mogą jak gdyby nigdy nic zatrudniać nadal na śmieciówkach. Z tym trzeba po prostu skończyć. Piszecie państwo w tej ustawie, że jej celem jest przywrócenie rentowności firm. To jest za mało. Te cele muszą być zdecydowanie ambitniejsze. Tym celem musi być odtworzenie dobrej jakości miejsc pracy. I to jest jedyny powód, dla którego w ogóle możemy rozmawiać w tej Izbie o wspieraniu prywatnych biznesów z publicznych pieniędzy. Bo przypominam, że te pieniądze pochodzą w większości z podatków, które płacą w Polsce pracownicy, i trzeba gospodarować nimi tak, żeby wynikła z tego korzyść była korzyścią całego społeczeństwa, a nie tylko wąskiej grupy właścicieli. Od kilku tygodni pan premier Morawiecki zaczął powtarzać po Lewicy, że pomoc państwa nie powinna trafiać do firm z rajów podatkowych. Bardzo dobrze, panie premierze. A teraz czas opanować kolejną lekcję. Pomoc państwa nie może się rozpłynąć w przepastnych kieszeniach nielicznej grupy prezesów firm. Ta ustawa wymaga poprawek, po to żeby zabezpieczyć interes publiczny. Dlatego Lewica opowiada się za skierowaniem jej do dalszych prac w komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 chciałbym przedstawić nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przedmiotowa ustawa jest elementem realizacji rządowego programu mającego na celu umożliwienie wsparcia ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach zmagających się z problemami finansowymi. Przyspieszone prace legislacyjne nad tą ustawą nie były wynikiem aktualnego kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią i związanego z nim wzrostu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, lecz sytuacją związaną z epidemią. Natomiast są trzy zasadnicze uwagi, które mamy, jeśli chodzi o ten projekt. Po pierwsze, dlaczego tak późno? Pani minister Emilewicz podczas wielu debat jeszcze poprzedzających tzw. pierwszą tarczę antykryzysową wspominała już o tym projekcie blisko 2 miesiące temu. Po drugie, wydaje się, że z dobrodziejstw tej ustawy wielu prowadzących działalność gospodarczą nie skorzysta. Ja jestem człowiekiem dużej wiary, ale mimo to nie sądzę, aby prowadzący zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, małe sklepy, sklepiki, którzy popadną w problemy w związku z obecną sytuacją, byli w stanie przebrnąć przez gąszcz wymogów biurokracji, który zawiera niestety ta ustawa. I po trzecie, powtórzę już za przedmówcami, te środki, które państwo przewidujecie, to jest kropla w morzu potrzeb, która absolutnie nie będzie miała jakiegokolwiek istotnego znaczenia, chodzi o pomoc w wyjściu z trudnych sytuacji, w których niewątpliwie wielu przedsiębiorców się znajdzie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja, jaka jest potrzeba chwili, choć doświadczenia obu ustaw, tzw. antykryzysowych, niestety nie pozostawiają dobrych wrażeń, nadziei na to, abyśmy mogli wspólnie coś w tej Izbie przygotować w atmosferze faktycznej, a nie tylko deklarowanej współpracy.

I na ten moment nasz klub będzie w tych dalszych pracach uczestniczył. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja przedstawi pan poseł Michał Urbaniak. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Otóż mam możliwość przedstawienia stanowiska koła Konfederacja w sprawie projektu o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Otóż ten rządowy projekt to w zasadzie kolejny ochraniacz dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przychodzi mi na myśl - już tak na wstępie - pewien wiersz. Mówię tu o wierszu Jana Kochanowskiego „Pieśń o spustoszeniu Podola”, a konkretnie chodzi o jego dwa wersy: „Nową przypowieść Polak sobie kupi, / Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. A już tłumaczę dlaczego. Otóż szanowna strono rządowa, proponujecie w tym projekcie szereg instrumentów dla firm, które de facto już mają przesłanki tego, że są w stanie upadłości. Proponujecie rozwiązania obwarowane szeregiem założeń niemal niemożliwym do spełnienia.

Dopiero kryzys związany z COVID-19 zmusił was do tego, by wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Ten projekt dotyczy zasadniczo małych, średnich przedsiębiorstw. Oczywiście nie tylko. Zakłada pożyczki oprocentowane, a okres kredytowania wynosi od 6 miesięcy do maksymalnie 18.

To jest za krótki okres. 50% zabezpieczenia, jakie przy tych pożyczkach narzucacie, to w przypadku też jakichś małych firm może być problematyczne. Mówiliście, w projekcie zapisaliście też, że wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane w 30 dni, maksymalnie w 45 dni. W przypadku przedsiębiorców, którzy są w stanie prawie że upadłości, 45 dni to jest za dużo czasu. 14 dni - to mogłoby być akceptowalne w tym wypadku, bo to jest czas, w jakim firma jest w stanie jeszcze przeżyć. W innym przypadku koszty cały czas rosną, rosną zobowiązania, rosną też dzięki temu problemy. W tym projekcie zakładają państwo, że rocznie przeznaczycie na ten projekt 120 mln zł. 120 mln zł, ale trzeba wziąć pod uwagę to, ile obwarowań prawnych będzie przy składaniu wniosków i jak będzie wyglądać sytuacja z przygotowaniem planów restrukturyzacji.

Jeśli faktycznie Prawu i Sprawiedliwości, stronie rządowej też, zależy na tym, aby polskie firmy się rozwijały, aby ratować polską gospodarkę, to sami przedsiębiorcy mówią jasno o tym, co jest im dzisiaj potrzebne. To, co dzisiaj, w zasadzie już od miesięcy, jest przypominane, to choćby to, co wprowadziliście, czyli split payment. To nie jest zdrowy sposób ściągania podatków z przedsiębiorców. Blokujecie w ten sposób pieniądze, którymi przedsiębiorcy w ciągu miesiąca mogliby swobodnie obracać, a dopiero potem płacić podatek. W tej sytuacji split payment blokuje to. To są naprawdę wielkie, wielkie pieniądze, a ściągnięcie w przypadku nadpłaty pieniędzy z konta split payment graniczy z cudem.

Dopiero po transakcji to powinno się wydarzyć.

Apelujemy, żebyście tym się zajęli, a nie takim projektem, który jest zapchajdziurą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy oświadczenia w imieniu klubów i koła. Przechodzimy do pytań.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

O tym mówił tutaj Waldemar Sługocki występujący w imieniu Koalicji Obywatelskiej.

Mam takie pytanie: Czy państwo widzicie potrzebę specrozwiązań właśnie dla tej grupy, ponieważ to ona już dzisiaj praktycznie jest zagrożona tym, że lada moment przestanie działać, a wielu z nich już nie działa. To jest też pytanie o historię, jak się w ogóle przygotowywano do czasów kryzysowych, które zawsze przecież przychodzą. Może by brać przykład z samorządów, od marszałków województw, podam przykład marszałka województwa wielkopolskiego (Dzwonek), który kiedyś zdecydował o tym, że wprowadzono tzw. instrumenty zwrotne z wykorzystania środków europejskich i dzisiaj, proszę państwa, zadeklarował już ponad 70 mln zł, i to już jest do wzięcia, przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju na płynność bieżącą i na ratowanie przedsiębiorstw. To jest zdecydowanie za mało. Dobrze. Biurokracja jest tak duża przy tym projekcie, że na pewno w trakcie prac w komisji będziemy dążyli do tego, żeby na specjalną sytuację - a jesteśmy w specjalnej sytuacji kryzysowej - przygotować rozwiązania bardzo proste, oczywiste i szybkie.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czytając tę ustawę, chciałoby się powiedzieć: Panie premierze, rządzie, panie ministrze, halo, tu Ziemia, tu wiosna 2020 r., tu czas pandemii i największego kryzysu ekonomicznego od lat. Z czasów, kiedy pan premier Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej premiera Donalda Tuska. Z czasów, których już nie ma, które bezpowrotnie minęły wraz z wybuchem epidemii. Trudna sytuacja, na którą w założeniu miała odpowiadać ta ustawa, to dziś nie przypadek, nie wyjątek dotyczący tylko niektórych przedsiębiorców. Dziś w trudnej sytuacji znajdują się setki tysięcy fryzjerek, kwiaciarek, hotelarzy, restauratorów, właścicieli sklepów, organizatorów imprez masowych, kosmetyczek, instruktorów. I oni wszyscy, ci wszyscy ludzie czekają dziś na adekwatne działania, na prawdziwy ratunek - nie przed przejściowymi trudnościami, ale przed realnym bankructwem. Moje pytanie brzmi zatem: Na co państwo czekają? Kiedy zajmiecie się ustawą, [[Dzwonek]] którą dała wam w tym kryzysie Lewica, o finansowaniu przez państwo kosztów stałych przedsiębiorstw? Dziękuję bardzo, pani poseł.

Pani Marszałek! Mam dwa pytania. Czy Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma realizować zadania wynikające z tej ustawy, jest przygotowana operacyjnie do wprowadzenia wejść kapitałowych? Drugie pytanie dotyczy samorządów, bo w przypadku ratowania przedsiębiorstw będzie to miało na pewno duży wpływ na wpływy z podatków do kas samorządów. Już dzisiaj samorządy wykonują bardzo dużo zadań za rząd. Nie idą w ślad za tym pieniądze. Pokrywają koszty pseudoreformy edukacyjnej. Dzisiaj samorządy wielokrotnie wspierają szpitale, przedsiębiorców, ratują lokalne firmy, natomiast ze strony rządu nie płyną żadne instrumenty, które miałyby pomóc samorządom. Czy w obliczu tego kryzysu, pomocy przedsiębiorcom, przewidujecie państwo również wsparcie samorządów?

Pan poseł Marcin Kulasek, klub Lewica.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pomoc dla przedsiębiorców powinna być, ale Lewica nigdy nie zgodzi się na bezwarunkowe pompowanie pieniędzy do biznesu. Firmy nie działają tylko dla dobrobytu menedżerów czy właścicieli, ale również po to, aby dawać ludziom dobrze płatną i bezpieczną pracę. Nie chcemy scenariusza, w którym firma dostanie pomoc od państwa, a pierwszą inwestycją będzie wymiana floty limuzyn dla zarządu. Ludzie to widzą, kłują ich w oczy takie inwestycje, rozmawiają o nich i krew ich zalewa, a w czasie kryzysu zalewa ich nawet bardziej niż zwykle.

Pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Projekt ustawy, który omawiamy, jest na normalne czasy. To nie jest projekt ustawy na stan kryzysu epidemicznego ani na stan nadzwyczajny, w jakim znajduje się polska gospodarka.

My tu nie mówimy o utracie konkurencyjności. Polskie przedsiębiorstwa są konkurencyjne, natomiast po prostu nie mogą funkcjonować ze względu na ograniczenia narzucone przez rząd, przez władzę. Jest potrzebna zupełnie inna ustawa. Dziwię się w ogóle, że 4 lata czekaliście z taką ustawą o pomocy publicznej, która mogła być wprowadzona już po 2016 r. - dlatego że były takie możliwości - i dopiero teraz, chcąc sprawić wrażenie, że dajecie Polakom jeszcze jeden instrument pomocowy, wprowadzacie ten projekt ustawy. To jest zupełnie bezużyteczny projekt. On jest dobry, jak powiedziałem (Dzwonek), na dobre czasy, natomiast z całą pewnością nie pomaga gospodarce. Chciałem was zapytać na koniec, panie ministrze, jakie macie jeszcze możliwości finansowe. Wiemy, jaki jest deficyt w obecnym budżecie, i wiemy też, jaka jest skala potrzeb pożyczkowych, 78 mld pożyczone od NBP. Pani poseł Monika Pawłowska, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pytam, czy rząd w końcu zajmie się problemem lotniska w Świdniku. Spółka Port Lotniczy Lublin SA, na którą ani minister Sasin, ani minister Soboń nie zwrócili uwagi, to lotnisko regionalne, na którym zbijacie kapitał polityczny, a teraz nie macie za grosz przyzwoitości, aby odpowiedzieć na apel o pomoc. To jest właśnie wasza polityka. Nie ma koronawirusa, chwalicie się osiągnięciami. Jest koronawirus, nie potraficie wziąć na siebie odpowiedzialności. Port Lotniczy Lublin SA woła o pomoc, bo został pominięty przez wasz rząd. To wasza wina, że tego nie dopilnowaliście. Zajmujecie się drukowaniem kopert, a nie możecie zająć się ratowaniem m.in. motoru województwa lubelskiego, z którego i wy korzystacie. Nie ma nic prostszego w tym momencie niż zagłosowanie za poprawką Lewicy. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie ministrze, nie będę powtarzał już krytycznych uwag, aczkolwiek mam nadzieję, że gros z nich uwzględnicie państwo być może w przyszłości. 120 mln rocznie chcecie państwo przeznaczyć na realizację tejże ustawy. Panie ministrze, czy nie lepiej byłoby, nie korzystniej z punktu widzenia potrzeb polskich przedsiębiorców, aby te alokacje roczne były nieco inne, czyli żeby w roku 2020 był zdecydowanie największy poziom finansowania, w 2021 r. - nieco mniejszy i każdego roku mniejszy? Dlatego że dzisiaj potrzeby przedsiębiorców są zdecydowanie największe.

Pani poseł Marta Golbik, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 45 dni - a w najgorszym wypadku, przy odwołaniu, ponad 100 dni - oczekiwania na decyzję. Przecież każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej, wie, że w tej sytuacji większość firm po prostu padnie.

Tak naprawdę powinniśmy się zająć dzisiaj jedną rzeczą: zacząć ufać przedsiębiorcom i realnie patrzeć na ich potrzeby. Dlaczego w innych krajach to może działać na zasadzie oświadczenia? Dlaczego pieniądze mogą przychodzić natychmiast, a u nas przedsiębiorcy muszą czekać kilkadziesiąt dni, czasem ponad 100 dni na to, żeby dostać jakąkolwiek pomoc? Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie wierzę w ten projekt. Nie wierzę, bo, po pierwsze, jest późno, po drugie, jest trudny, po trzecie, jest mało środków finansowych, a po czwarte, o czym powiedział pan prof. Rosati, to nie ten czas. Proszę państwa, w ciągu miesiąca trzeci raz debatujemy nad trzecią tarczą.

Rząd niezwykle pięknie mówi, ale prawda jest inna. Jest prawda rządowa i jest ta prawda, kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami - to zupełnie inaczej wygląda. Panie premierze, jeśli mogę coś [[Dzwonek]] doradzić: mniej konferencji prasowych, więcej pieniędzy. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Wejścia kapitałowe nie oznaczają nic innego jak objęcie przez Skarb Państwa obligacji, akcji lub udziałów przy podwyższeniu kapitału zakładowego ratowanych przedsiębiorstw. Wysoka Izbo, drodzy państwo, takie działania można nazwać próbą nacjonalizacji przedsiębiorstw. Parlament powinien mieć silniejszy mandat w zakresie nadzoru nad tymi działaniami. Niezwłocznie należy przygotować taki nadzór, aby przedstawiciele społeczeństwa mieli możliwość kontroli nad udzielonym wsparciem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Na koniec pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia postojowego, czekają już ponad miesiąc. Jeśli ta ustawa ma działać dokładnie tak samo, to nikogo nie uratujecie. To jest tylko i wyłącznie po to, żebyście przed kamerami pokazali, że chcecie ratować, że macie pomysł, a to, że nie uratujecie nikogo, już mało kogo będzie interesowało. Dziękuję bardzo, panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania pań i panów posłów odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju minister Krzysztof Mazur. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mówiłem o tym na samym początku i państwo doskonale o tym wiecie, że tak naprawdę to jest ustawa nie na ten moment, tylko na kolejne 10 lat.

Jeżeli stwierdził pan, panie pośle Zandberg, że mówimy także o wejściu kapitałowym państwa, to tak, tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, która dzisiaj ruszyła o godz. 18, jak powiedziałem, dokładnie to zakłada. Tak więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że to jest jedyne działanie i że tak długo czekaliśmy na tę ustawę, bo to jest, jak policzyłem, szósta ustawa: trzy COVID-owe, czwarta była o dopłacie do kredytu, piąta była o instytucjach rozwoju. Także argument, panie pośle Sługocki, dotyczący czasu, jest absolutnie nieprawdziwy.

Okej, ale pamiętam czasy SLD, pamiętam czasy Platformy. Nie pamiętam, żeby w ciągu 14 dni taki proces tak szybko działał. Po drugie, jeżeli mówimy o barierach administracyjnych, to rzeczywiście bardzo chętnie w komisji popracujemy nad tym, żeby było ich jak najmniej. Jak już nie będzie takiego szerokiego audytorium, to pokażemy państwu, jakie są wytyczne Komisji Europejskiej. Jutro mamy kolejne spotkanie z nimi i dyskutujemy z nimi na temat tego, dlaczego te wytyczne akurat do tej podstawy, która nie jest podstawą COVID-ową, jak powiedziałem, jest inną podstawą, sprzed czasów COVID.

Co jest najśmieszniejsze? Nie jest prawdą, panie pośle Sługocki, że tutaj, w tej ustawie, są środki europejskie. To są środki polskie, z polskiego budżetu, natomiast są oparte na wytycznych Komisji Europejskiej. To jest najciekawsze, że tak naprawdę własnych środków nie możemy wydawać tak elastycznie, jak byśmy chcieli.

Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby to było jak najprostsze, ale gdy na posiedzeniu komisji przedstawimy wytyczne Komisji, to sami zrozumiecie, na czym polega kłopot. Panie Pośle Zandberg! Mówi pan o tym, że kapitał wchodzi do firm. Chcę zwrócić pana uwagę na to, że właśnie dzisiaj ten mechanizm tarczy finansowej, 25 mld dla tych największych firm, to jest właśnie ten mechanizm. Jeżeli mówicie, że te 150 mln, 120 mln plus 50 mln to jest za mało, dzisiaj uruchomiliśmy PFR dla dużych firm w wysokości 25 mld. I tam także jest opcja wchodzenia kapitałowego państwa do firm.

Tak, bo to jest skala na restrukturyzację już po COVID. Co do kwestii działalności ludzi, że to ma iść na działalność ludzi, a nie prezesów, absolutnie, zgadzam się z wrażliwością Lewicy. I wiecie doskonale, że środki w ramach tej ustawy będą przyznawane w oparciu o szczegółowy plan restrukturyzacyjny. Jeśli w tym szczegółowym planie restrukturyzacyjnym nie będzie ani złotówki na flotę samochodową, nie będzie takiej możliwości. Znowu rozmawiamy o jakiejś fantasmagorii. To jest też bardzo ciekawe, bo z jednej strony mówicie: ma być mało wniosków, mało papierologii, ale z drugiej strony: ma pójść na to, a nie na tamto. Administracja działa w ten sposób, że jeżeli ma plan restrukturyzacji, to wie, że może przypilnować, że pójdzie na plan restrukturyzacji, a nie na flotę, tak że tutaj też jest pewna niekonsekwencja. Jeśli chodzi o kwestię dni - 14 czy 30 - chętnie w komisji przyjmiemy te poprawki. Chcielibyśmy, żeby to było w ciągu 1 dnia albo 2 dni, natomiast zobaczycie, czy to jest możliwe, w oparciu o te wytyczne Komisji. Jeśli chodzi o zawieszanie kar, padł taki postulat, bodajże pani poseł Urbaniak. Tarcza pierwsza i druga zakłada zawieszanie kar, a zatem mówimy o prawie, które już przez tę Izbę przeszło. Tak że prosiłbym, żeby nie postulować rzeczy, które już przeszły. Jeżeli chodzi o kwestię ARP, czy jest przygotowana. Tak, jest dobrze przygotowana. Mówiłem o tradycji tej instytucji. Tak, ma już podobny program, kilka podobnych programów na swoim koncie, tak że wydaje się nam, że ARP jest do tego dobrą instytucją. Jeżeli chodzi o kwestię samorządu, to również wiecie doskonale, że w tarczy 3.0 są rozwiązania dla samorządu, tak że wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądała stabilność budżetowa samorządów, odsyłam do tego aktu prawnego. Jeżeli chodzi o kwestie. Uwagi do pana posła Rosatiego także przekazałem. Mamy nadzieję, że będziemy już poza epidemią. I tak potrzebujemy szczegółowych planów restrukturyzacyjnych dla firm w tym kontekście. Jeżeli chodzi o lotnisko w Świdniku, bardzo proszę o pytanie na piśmie.

Czy jeszcze coś? Chyba o nacjonalizacji padło kilka słów, więc mogę odpowiedzieć tylko tak. Przez tę Izbę przeszła tarcza 1.0, która dawała możliwość kapitałowego zaangażowania, m.in. Polskiego Funduszu Rozwoju, i w ramach tego jest uruchomiona tarcza finansowa, która daje możliwość wchodzenia kapitałowego państwa, jeżeli chodzi o wsparcie firm. Mamy konkretne firmy, które stają, nawet na konferencji prasowej, jak państwo widzicie, z panem premierem, i tak, oczekują tego, że na czas kryzysu państwo pomoże także w ten sposób, że obejmie część akcji w taki sposób, żeby dokapitalizować te przedsiębiorstwa, żeby one uzyskały płynność. Tak że jeśli przez ograniczenia czasowe, bo już przekroczyłem 3 minuty, nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, bardzo proszę o złożenie pytań na piśmie i o pracę w komisjach. Jestem otwarty na to.

Dziękuję bardzo.

Nie powiedziałem, że pomoc publiczna pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, tylko powiedziałem, że stosowne rozporządzenia Unii Europejskiej umożliwiają przekazywanie środków publicznych krajowych na poczet polskich podmiotów gospodarczych.

Tak czy nie? Proszę odpowiedzieć. Jeszcze pan minister prosił o głos. 30 sekund. Był pan łaskaw powiedzieć, że w narracji pana premiera Morawieckiego jest pewna niespójność, ponieważ krytykuje Unię Europejską, a zarazem korzysta z narzędzi Unii Europejskiej. Mogę powiedzieć, panie pośle? A więc na przykładzie tej ustawy widać wyraźnie, że obostrzenia, które funkcjonują w Unii Europejskiej, które nie pozwalają na pomoc publiczną firmom nawet z budżetu krajowego. Przepraszam, tylko dokończę.

Mówiono, że potrzebujemy zniesienia capu dla pomocy publicznej, dlatego że jest ona zbyt sztywna i nie pomaga nam reagować.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zawarty w druku nr 300, do Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.